Ten fundusz dobrze sprawdzał się przez lata w obszarze sportu, wsparcia przez. Jest to kolejny instrument, jeden z funduszy, którym dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Filozofią było to, iż na specjalnie wydzielony rachunek będący w dyspozycji ministra sportu trafiały środki z opłat w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług od przedsiębiorców świadczących usługi będące reklamą napojów alkoholowych. Taka to konstrukcja została przyjęta.

W związku z tym dobrze, że po latach w wyniku analizy dokonujemy pewnej zmiany, polegającej na tym, że owszem, dyspozycja nie pozostaje dotknięta, bo zgodnie z ideą to minister właściwy w obszarze sportu będzie dysponował tymi pieniędzmi, natomiast sprawę.

W związku z tym my, jeśli chodzi o te nowelizowane przepisy, jako Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska nie zgłaszamy żadnych poprawek. Sprawozdanie niewiele różni się od tego przedłożenia rządowego, myśmy tylko wyregulowali pewne kwestie legislacyjne, redakcyjne. W imieniu moich koleżanek i kolegów z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska wnioskuję, abyśmy przyjęli tę nowelizację. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Janusza Szopińskiego z klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi utworzony został Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym, a jego przychody są wpływami z tytułu opłat, które podmioty świadczące usługi będące reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Realizacja zajęć sportowych dla uczniów naszych, polskich szkół wspierana jest przez ten fundusz od roku 2003.

Natomiast w roku 2009 przyjęto priorytet programowy, którym była nauka pływania. Przedmiotowe rozwiązanie miało na celu upowszechnianie umiejętności pływania oraz niwelowanie barier w dostępie do zorganizowanych form aktywności fizycznej poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w ogólnopolskich programach upowszechniania nauki pływania pod nazwą „Umiem pływać”

Z satysfakcją chciałbym powiedzieć, że od początku prac nad uchwaleniem tej ustawy, ustawy dobrej dla rozwoju polskiego sportu, ustawy dobrej dla młodzieży, ustawy dobrej dla dzieci, obecny był rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecni byli posłowie, którzy wtedy zasiadali tutaj w tych ławach poselskich, m.in. pan poseł Tadeusz Tomaszewski, który z tego miejsca przemawiał w imieniu komisji kultury fizycznej i polecał Wysokiej Izbie przyjęcie rozwiązań w tej ustawie.

Chodzi o to, aby zmiany legislacyjne mogły zoptymalizować system poboru opłat i skuteczność wywiązywania się przez podatników z obowiązków nałożonych ustawą o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To jest dobry projekt. Klub Lewica będzie głosował za przyjęciem rozwiązań przedstawionych w tym projekcie. Projekt ten otrzymał również stosowne dobre opinie zarówno Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, co mój klub przyjmuje z dużym uznaniem. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Dariusza Kurzawę, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Europejskich Demokratów, Konserwatystów mam zaszczyt zaopiniować zmiany w ustawie o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odpowiednio druki nr 209 i 703. W obecnym stanie prawnym inny podmiot otrzymuje opłatę należną z tytułu reklam napojów alkoholowych, a do innego składa się deklarację. Wpływa to niekorzystnie na efektywność systemu poboru opłat.

Wobec tego w ocenie klubu Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Europejskich Demokratów, Konserwatystów wprowadzenie proponowanych zmian, tzn. scedowanie na urzędy skarbowe wszystkich czynności związanych z poborem opłat i składaniem deklaracji, jest właściwe. Wprowadzenie e-deklaracji oraz doprecyzowanie systemu egzekucji należności również wpłynie pozytywnie na realizację zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Mój klub Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści pozytywnie opiniuje przedstawione przez komisję projekty zmian.

Dziękuję bardzo. Zapraszam pana posła Krzysztofa Tuduja, Koło Poselskie Konfederacja. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jestem jak najbardziej za promocją sportu, za aktywnością sportową młodych ludzi, szczególnie w obecnych smartfonowych czasach. Ale jeśli pochylamy się nad problemem alkoholowym, to sport nie jest pełną i jedyną odpowiedzią. Równie dobrze można organizować zajęcia z tego, jak trenować silną wolę, wyznaczać w życiu cele. Można też dawać realne ostrzeżenie: unaoczniać, poprzez uczestnictwo w sesjach grup wsparcia dedykowanych anonimowym alkoholikom, do czego może prowadzić używanie alkoholu jako substancji psychoaktywnej. Trzeba mocno podkreślić, że nie nakazy i rozkazy stanowią o wychowaniu w trzeźwości, tylko przykład.

Taka metoda zwalczania problemu alkoholowego jest długofalowo nieskuteczna. Stanowi tylko sposób na uśpienie wyrzutów sumienia, daje ustawodawcy i urzędnikom poczucie, że coś tam się robi, że czemuś się przeciwdziała. Trzeba promować wiedzę wśród dorosłych Polaków, aby korzystali z alkoholu z umiarem. Jak? Może przy użyciu telewizji publicznej, po to ona chyba istnieje.

Należałoby kierować je bezpośrednio do osób, które są w grupie ryzyka, aby życiowym doradcą nie stała się spotykana codziennie flaszka czy też ciągle przerażająco modna flaszeczka małpeczka. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która jest nowelizowana omawianym projektem, została uchwalona w 1982 r., więc jeszcze w cieniu stanu wojennego. Od tamtego czasu była wielokrotnie nowelizowana.

Może w ogóle warto skończyć nowelizację i spojrzeć na ten problem w sposób świeży, z uwzględnieniem badań prowadzonych w tym milenium i obecnej wiedzy, przygotować po prostu nową ustawę. Na koniec trzeba powiedzieć, że nie mamy jeszcze badań na temat spożycia alkoholu w 2020 r. Powtarzane zatrzymanie gospodarki, nieumiejętnie prowadzona polityka informacyjna na temat walki z COVID-em prawdopodobnie doprowadzą również do wyższego spożycia alkoholu w tym roku. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie wiem, czy państwo wiedzą, że powstała ona dlatego, że gen. Jaruzelski był abstynentem. Rzeczywiście cała ta ustawa nadaje się do kosza. Ma szereg bardzo szkodliwych zapisów. Zamiast zlikwidować te zapisy, państwo zajmują się jakimiś nieistotnymi szczegółami. A jednym z bardziej szkodliwych zapisów tej ustawy jest jedyny w Europie zapis zakazujący sprzedaży alkoholu przez Internet. To zapis absurdalny, uderzający w polską gospodarkę, w polskich producentów czy to piwa regionalnego, rzemieślniczego, browarów kontraktowych, czy też innych napojów.

Stan zatrudnienia został już zredukowany o prawie 70%.

Uwaga: Jak to obchodzą wielkie sieci, inne firmy? Tak to się odbywa. Na tym posiedzeniu Sejmu będzie taka poprawka. Apeluję do wszystkich posłów, by wreszcie wyrzucić ten szkodliwy przepis z tej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Nie wiem, czy posłowie Lewicy zagłosowali niewłaściwie. Zapraszam panią poseł Joannę Fabisiak z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska.

Pan poseł Suchoń jak zwykle jest, więc proszę bardzo. Panie Marszałku! Cieszę się, że pan marszałek z taką radością powitał mnie na tej mównicy, ale też, jak myślę, temat jest. Ale gdzież mi do pana marszałka tutaj, w tej Izbie. Panie marszałku, kto jak nie my wzajemnie powinniśmy sobie te komplementy prawić, prawda? A że temat jest istotny i sprzyjający, powiedziałbym, temu, o czym wszyscy marzymy, czyli zdrowiu publicznemu, chciałem zapytać panią minister, korzystając z okazji, że ta ustawa jest procedowana, o to, w jaki sposób w tym roku zostały wykorzystane środki z tego funduszu, ponieważ trudno na stronach internetowych ministerstwa znaleźć informacje dotyczącą konkursów. Są informacje z poprzednich lat, natomiast tegorocznych ja przynajmniej nie mogłem znaleźć, więc bardzo bym prosił o te informacje.

Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do właściwego ministra, który jest dysponentem środków na realizację zadań sportowych w kontekście Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Pytam o to z powodu raportu Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, iż zmalał odsetek dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat, podejmujących aktywność fizyczną zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Myślę tutaj o 60 min aktywności dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Jak to się ma do planowanych (Dzwonek) przez jednostki samorządowe inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej? Myślę tutaj np. o pierwszym w powiecie sępoleńskim basenie w Sępólnie Krajeńskim, o inwestycjach dotyczących obiektów sportowych w Bydgoszczy: basenu rehabilitacyjnego czy budowy hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią poseł Zofię Czernow z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Pani Minister! Ja chciałam zapytać o fundusz. Jak państwo szacują, jakie będą roczne przychody tego funduszu po uwzględnieniu zmian, które są w tej chwili procedowane? To pierwsze pytanie. Ile z tych pieniędzy otrzymują szkolne kluby sportowe? Czy w ogóle otrzymują? Tych pieniędzy w klubach brakuje, i to bardzo.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Tomasz Olichwer, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Zapraszam, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rząd zmienia ustawę w kwestiach mało istotnych ze względu na sam problem zdrowotny osób uzależnionych i jakość życia ich rodzin. Jak widać, do tej pory nie widzi potrzeby wprowadzenia przepisu o przymusowym leczeniu osób uzależnionych, który jest wyłącznie stosowany w przypadku zagrożenia życia lub utraty zdrowia. Moim zdaniem jest to bardzo istotna kwestia. Nadal nie dostrzegacie państwo tragedii rodzin, żon, matek i dzieci osób uzależnionych, nie widzicie potrzeby udzielenia im prawdziwej pomocy, zarówno krzywdzonym, jak i osobie bezpośrednio uzależnionej. Warto podkreślić, że osoba uzależniona nie jest w stanie racjonalnie decydować o swoim losie, dlatego w takim przypadku przymus oznacza jedyny ratunek. Obecne prawo tylko przykrywa i głaszcze ten problem, a rodziny żyjące na co dzień z osobą uzależnioną są często bite, zastraszane, nie mają środków finansowych na życie, [[Dzwonek]] nie mają się gdzie wyprowadzić i nie mogą zgłosić takiej osoby na przymusowe leczenie. Czy to jest pomoc? Odpowiedzcie sobie państwo sami. Tak - dla Unii, nie - dla weta. Dziękuję serdecznie. Będziemy się łączyli z panią posłanką Katarzyną Kretkowską.

Problem alkoholowy w Polsce jest jednym z największych problemów społecznych - mamy 2% alkoholików i 12% nadużywających alkoholu. Służba zdrowia jest obciążona leczeniem samego alkoholizmu i chorób współistniejących. W związku z tym mam pytanie do rządu: Czy nie należałoby jednak ograniczyć reklamy alkoholu, mimo że ona już jest ograniczona np. w telewizji do późnowieczornych godzin nocnych, ograniczyć te reklamy (Dzwonek), a finansować sport dzieci i młodzieży z budżetu państwa? Byłoby to i tańsze - tak sądzę, biorąc pod uwagę środki, jakie wydaje służba zdrowia na leczenie alkoholizmu - i lepsze dla całego społeczeństwa, dla osób, które mają problem, i dla ich rodzin. Dziękuję. Pan poseł Paweł Papke, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Projektowane zmiany legislacyjne mają na celu zoptymalizowanie systemu poboru opłat i podniesienie skuteczności wywiązywania się podatników z obowiązków nałożonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Aktualne uwarunkowania powodują, że inny podmiot otrzymuje należną opłatę, a inny deklarację, co niekorzystnie wpływa na efektywność systemu poboru opłat. Stąd moje pytania. Czy doprecyzowanie przepisów tej nowelizacji odnoszących się do opłaty będzie prowadzić do wszczynania zaległych postępowań windykacyjnych wobec przedsiębiorstw i tym samym ściągnięcia należności na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów? Do tej pory mieliśmy bowiem problem z efektywnością systemu poboru opłat i nie wszystkie należności znalazły się na rachunku. I drugie pytanie, oczywiście: Ile według szacunków ministerstwa wynoszą zaległości podatkowe, które nie są opłacone? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Jakub Rutnicki, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Proszę. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Pokazujemy te rzeczy.

Myślę, że mogłoby to być bardzo skuteczne. Pan poseł Jan Szopiński, Klub Parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż tak. W tym czasie z przyczyn bliżej nieznanych w tempie olimpijskim rząd zmienił ustawę o działach administracji rządowej. I nie byłoby tu żadnych wątpliwości, tylko że w tej ustawie o działach administracji rządowej wprowadził rewolucyjne zmiany w zakresie administrowania polskim sportem, współpracy ze związkami sportowymi i finansowania polskiego sportu. Tempo olimpijskie było takie, że nie mając ustawy, premier w październiku br. powołał pełnomocnika do spraw funkcjonowania Narodowego Centrum Sportu.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Artur Dziambor z koła Konfederacji. Już w dobrym zdrowiu, jak widzę, na szczęście. Wysoka Izbo! Każdy z nas ma jakieś swoje używki. Dla niektórych są to papierosy, dla niektórych jest to alkohol, dla innych jest to szybka jazda samochodem, dla jeszcze innych jest to cukier, dla mnie pizza, dla jeszcze innych miękkie narkotyki, które w sumie nie wiadomo dlaczego są u nas nielegalne.

Państwo nie powinno w tym w ogóle uczestniczyć, a podatki, które płacimy, powinny być odpowiednio celowe. Powinniśmy wiedzieć, ile z naszych podatków i w jakim stopniu wspiera walkę z alkoholizmem, którą - tak jak powiedziałem - powinni się zajmować inni, nie państwo, walkę z innymi używkami i ile z naszych podatków idzie na promocję sportu. Promocję sportu, czyli w ogóle sport, który również powinien być (Dzwonek) całkowicie wyłączony z państwowego budżetu, bo to nie państwo powinno się sportem zajmować. Dziękuję bardzo i dziękuję za pozwolenie na przedłużenie wypowiedzi. Proszę bardzo, byłem zainteresowany katalogiem pokus, które pan wymienił, bo to różnie z nimi bywa. Pani poseł Magdalena Łośko, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dotychczas obowiązujące przepisy stanowiły, że 10-procentowa opłata za usługi będące reklamą napojów alkoholowych zasilała bezpośrednio rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, oczywiście z przeznaczeniem na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Pytanie: Czy wprowadzenie bezpośrednio pośrednictwa urzędów skarbowych w przekazywaniu środków na rachunek ministra do spraw kultury fizycznej będzie się wiązało z kosztami i uszczupleniem środków na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów? Dziękuję serdecznie. Tak myślę o panu pośle Arturze Dziamborze. Wie pan, jak ministrowie PiS-u do nas stoją tyłem, to się dobrze nie czujemy. Proszę, Wiesław Buż, poseł klubu parlamentarnego Lewica. Wiem, jestem z tego znany. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projektowana ustawa zakłada, że zmiany nie wpływają na wydatki budżetu państwa i samorządu. Moim zdaniem wpływają, bo wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w chwili obecnej środki te trafiały do właściwego ministerstwa, w tym wypadku ministerstwa kultury fizycznej. Obecnie po przyjęciu tej ustawy będą trafiać na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Czy oprócz bezpośredniego przekonania, że tych środków dla uczniów... bezpośredniego przekazania tych środków dla uczniów będzie więcej, czy zwiększy się wysokość wpłat na fundusz zajęć? Bo, powiedzmy, nie będzie algorytmu ani podziału. Nie wierzę również w to, że do tej pory wszystkie środki trafiały z powrotem do uczniów, bo też nie ma o tym mowy w żadnych sprawozdaniach. Ile dostawało środków ministerstwo? Dziękuję serdecznie, panie pośle. Na te pytania postara się odpowiedzieć sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu pani minister Anna Krupka. Zapraszam, pani minister.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przede wszystkim zacznę od tego, że opłaty za reklamę, wynikające także z tej ustawy, dzisiaj są przeznaczane na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów. W tym roku, bo padały tu takie pytania, finansowaliśmy z niej choćby takie akcje i programy jak „Umiem Pływać”, programy dotyczące upowszechniania sportów zimowych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

W przyszłym będzie to ok. 21 mln zł, natomiast zmniejszenie środków na 2021 r. wynika z wykorzystanych już środków z okresów poprzednich. Natomiast przychody z opłaty za reklamę planowane są na tym samym poziomie.

Więc de facto na ten cel w przyszłym roku przeznaczymy więcej.

Właściwi w sprawie opłaty za reklamy napojów alkoholowych będą naczelnicy urzędów skarbowych, a aktualna kwota należności wymagalnych wraz z odsetkami to ok. 100 tys. zł. Dysponentem Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów jest i będzie minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Padało tu pytanie o kluby sportowe. Otóż chciałam podkreślić, że takie stwierdzenie jest absolutnie nieuprawnione. W tym roku przeznaczyliśmy na małe i średnie kluby sportowe w ramach rządowego programu „Klub”, który utworzyliśmy w 2016 r., ok. 55 mln i wszelkie wnioski, które zostały złożone przez kluby zgodnie z wymogami formalnymi, były dofinansowywane, czyli każdy klub, który złożył poprawny wniosek, otrzymywał wsparcie. Tych klubów było... 4902 kluby otrzymały wsparcie. To także wynikało z tego, że jest to wyjątkowy rok epidemii koronawirusa, a jednocześnie była rekordowa liczba klubów, które zostały objęte wsparciem. Nigdy nie było tak szerokiego wsparcia dla klubów sportowych. Któraś z pań posłanek wskazała także, że jej zdaniem aktywność fizyczna Polaków spada. Otóż z badań biura ministra w Ministerstwie Sportu wynika, że ta aktywność rośnie. Przytoczę choćby fragment tych wyników. Odsetek Polaków uprawiających aktywność fizyczną w czasie wolnym, bez chodzenia rekreacyjnego w wymiarze rekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia.

A więc ta aktywność wzrasta. Mam tu także inne dane, które to pokazują, i bardzo chętnie je udostępnię. Oczywiście my odpowiemy także na to pytanie na piśmie. Na resztę pytań, jeżeli na jakieś nie odpowiedziałam, także będziemy odpowiadać na piśmie. Dziękuję serdecznie, pani minister. Faktycznie, ja też obserwuję wzmożoną aktywność fizyczną Polek i Polaków. Bardzo często widać ich spacerujących. To idzie w dobrym kierunku moim zdaniem. A, jeszcze jest sprawozdawca. Miałem kartkę, że może pana nie być, panie pośle. A jakby pan myślał, że chciałem to zrobić złośliwie, to nie, nie. Chcę zauważyć do mikrofonu, że pan marszałek Terlecki jest bardzo dobrym wicemarszałkiem i mogę tylko. O, dziękuję za te oklaski. Panie pośle, jak pan pozwoli, bo nie będę z panem Terleckim wchodził w konflikt, ja też potwierdzam, że jest bardzo dobrym marszałkiem, aczkolwiek trochę innym.

Ja też chciałem podziękować pani minister i wszystkim członkom obu komisji za rzeczową dyskusję w tej ważnej sprawie i za zgodę, która panowała zresztą również i na tej sali. Dziękuję panu serdecznie. Już mogę zamknąć, tak? Patrzę na pana, który zawsze mnie kasuje złym wzrokiem. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej (druki nr 240 i 635) Proszę bardzo pana posła Wojciecha Zubowskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Łączymy się zdalnie. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Nie widzimy pana jeszcze. Proszę bardzo, panie pośle, zapraszam. Dzień dobry. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Połączone komisje, Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na posiedzeniu w dniu 24 września 2020 r. rozpatrzyły komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej, druk nr 240. Po dyskusji połączone komisje rekomendują przyjęcie załączonego projektu ustawy. Jako poseł sprawozdawca dodam od siebie, że projekt ten został przyjęty bez żadnego głosu sprzeciwu jakiegokolwiek posła biorącego udział w tymże posiedzeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Zapraszam pana posła Sławomira Zawiślaka, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W swoim wystąpieniu przedstawię stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej, druk sejmowy nr 240. Projektowana ustawa jest pozytywną reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na petycję skierowaną przez obywatela naszego kraju, którą to petycję komisja uznała za zasadną. Cieszy to, ponieważ dla nas wszystkich powinno być istotne wsłuchanie się w głos każdego obywatela i odniesienie się do jego wniosków, a szczególnie to odniesienie się pozytywne.

Celem ustawy jest dokonanie zmian w dwóch ustawach, ustawie o przedsiębiorstwach państwowych i ustawie o gospodarce komunalnej, w tym kierunku, żeby te zmiany dostosowały występujące w niej odniesienia i terminologię do aktualnego stanu prawnego wskazanego właśnie w petycji obywatelskiej. Zmiany te wynikają z przekształcenia Polskich Linii Lotniczych LOT, ale także wejścia w życie trzech ustaw: ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi obejmującej zakresem podmiotowym osoby wykonujące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych; ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; ustawy Kodeks spółek handlowych i oczywiście uchylenia ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym. Dotyczy kwestii zmiany przepisów w tych spółkach, tak jak powiedziałem, z życzeniem autora petycji. Te zmiany, tak jak powiedział poseł sprawozdawca, zostały pozytywnie zatwierdzone przez członków wymienionych przez posła sprawozdawcę dwóch komisji sejmowych. Ponieważ zasadniczym skutkiem społecznym i prawnym projektowanej ustawy będzie poprawa spójności i przejrzystości systemu prawnego, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proszę Wysoki Sejm o poparcie tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej przedstawić stanowisko odnośnie do projektu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej stanowiących reakcję na petycję obywatelską - o czym była tu mowa, za co dziękuję - wniesioną do Sejmu. Projekt ustawy należy określić jako projekt o charakterze technicznym, ujednolicającym, dostosowującym do stanu faktycznego istniejące ustawy.

W chwili obecnej zostały one zastąpione odpowiednio przez Kodeks spółek handlowych oraz Krajowy Rejestr Sądowy.

Jak wszyscy wiemy, Polskie Linie Lotnicze LOT są dzisiaj spółką prawa handlowego. Obydwie proponowane powyżej zmiany są zmianami dostosowującymi treść wskazanych ustaw do rzeczywistego stanu prawnego. Ich przyjęcie nie spowoduje jakichkolwiek daleko idących skutków prawnych. W art. 43 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych jest mowa o prawie do prowizji od zysku przedsiębiorstwa.

Ponadto w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych uchyla się art. 46 ust. 1b odnoszący się do uchylonej już i nieobowiązującej od 2001 r. ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.

Skutkiem tego projektowana ustawa ujednolica wysokość odprawy do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Analiza stanowiska Rady Ministrów co do przedłożonego projektu ustawy wskazuje, że art. 12 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi stanowi, iż może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność wynagrodzenia miesięcznego, natomiast przedłożony projekt określa sztywną wysokość w postaci odprawy równej 3-miesięcznemu wynagrodzeniu. W związku z tym klub Koalicji Obywatelskiej składa poprawkę w następującym brzmieniu: „W przypadku odwołania dyrektora przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność wynagrodzenia miesięcznego” Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pani poseł. Pan poseł Wiesław Buż, klub parlamentarny Lewica. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo!

Przedmiotowy projekt ustawy odnosi się wyłącznie do kwestii porządkowych i w intencji wnioskodawcy ma na celu dokonanie jedynie kosmetycznych zmian, i to tylko w tych dwóch ustawach. Dlatego uznać to należy za podejście wadliwe. Odnosząc się do zmian ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, należałoby się zastanowić, czy nie włączyć postanowień tej ustawy do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W jednym akcie prawnym powinny być skupione zagadnienia dotyczące majątku państwowego, np. w ustawie o aktywach państwowych. Wobec istniejącego rozproszenia licznych aktów prawnych odnoszących się do państwowych osób prawnych i agencji łatwo przeoczyć zapisy mówiące o tym, że w jednym podmiocie państwowym, gdzie wypłaty są ze środków publicznych, zarząd otrzymuje sześć odpraw, a w drugim 3-miesięczną odprawę. Te zapisy znajdują się w art. 1 pkt 2 proponowanej ustawy. Konkludując, technika legislacyjna zaproponowana w projekcie jest fragmentarycznym prostowaniem poszczególnych zagadnień, co powoduje, zamiast ucięcia problemu, mnożenie kolejnych drobnych zmian do ustawy. Podobne uwagi trzeba skierować co do fragmentu projektu odnoszącego się do ustawy o gospodarce komunalnej. Tu także autorzy czy autor projektu zaproponowali poprawki redakcyjne odnoszące się do zmiany nomenklatury obecnie obowiązujących ustaw, natomiast bardziej pilnym problemem, zdaje się, jest jednoznaczne uregulowanie standardów, według których obecnie działają spółki komunalne. W wielu przypadkach przestały one wykonywać zadania własne i ich przychody z działalności komercyjnej są wyższe niż z działalności na rzecz właściciela, najczęściej jednostki samorządu terytorialnego. Pozostał enigmatyczny zapis w art. 10 ustawy, który mówi o przystępowaniu do spółek działających poza strefą użyteczności publicznej albo tworzeniu spółek zajmujących się inną działalnością niż użyteczność publiczna. Brakuje zapisów odnoszących się do sytuacji, gdy dana spółka komunalna zajmuje się zarówno użytecznością publiczną, jak i inną działalnością - komercyjną. Ponadto zapis w art. 10 ust. 1 pkt 1 mówi o niezaspokojonych potrzebach na rynku lokalnym. Pojawia się więc pytanie, co to jest rynek lokalny. Czy chodzi o rynek lokalny dla siedziby spółki, czy rynek lokalny, gdzie są niezaspokojone potrzeby? Przykład: spółka komunalna z gminy A wykonuje na rzecz podmiotów z gminy B działalność komercyjną. Czy może? Czy rynek lokalny w rozumieniu przepisu odnosi się tylko do rynku obejmującego granice administracyjne gminy, która utworzyła spółkę, czy nie? Podsumowując, przedłożony projekt ustawy należy ocenić jako niekompletny z punktu widzenia potrzeby kompleksowych rozwiązań prawnych odnoszących się do funkcjonowania państwowych osób prawnych oraz spółek komunalnych. Projektowane rozwiązania, których celem jest usystematyzowanie nomenklatury dotychczasowych przepisów, same w sobie nie są wadliwe, jednak nie odpowiadają na problem jednoznacznego uregulowania standardów, w jakich obecnie działają spółki komunalne i państwowe osoby prawne. Projekt został złożony jako petycja zgłoszona przez uprawniony podmiot w interesie publicznym. Parlamentarny klub Lewicy da poparcie tej regulacji, ale jednoznacznie zwracam uwagę na fakt, że to minister Sasin powinien wziąć się do roboty i rozpocząć pracę swojego resortu na rzecz dopasowania istniejącego prawa do nowych warunków, które powstały chociażby w wyniku powołania nowego ministerstwa, Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jednocześnie chciałem serdecznie podziękować za złożenie petycji oraz inicjatywę i pracę na rzecz zmiany oraz poprawy istniejących niedoskonałości w polskim prawodawstwie w obrębie przedsiębiorstw państwowych i spółek komunalnych. Dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Mieczysława Kasprzaka z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści, jest to duży klub w tej chwili, zrzeszający szereg podmiotów, chcę zabrać głos w sprawie procedowanej ustawy z druku nr 240 i sprawozdania z druku nr 635.

My często, a w tej chwili - bardzo często, zmieniamy podporządkowanie firm, instytucji, gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa, czasami nawet kilkakrotnie w przeciągu jednej kadencji parlamentarnej, w zależności od tego, jakie pomysły ma rząd.

Dlatego powinniśmy tego przestrzegać. Oczywiście nasz klub poprze te rozwiązania, bo one są logiczne, normalne, tylko powinniśmy się wystrzegać takich sytuacji, że to wychodzi nie od ustawodawcy.

Pan poseł Michał Urbaniak, koło Konfederacja. Zapraszam uprzejmie, panie pośle.

Panie Marszałku! Co do propozycji zmiany ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej zasadniczo nie mam większych zastrzeżeń. To jest prosta, kosmetyczna ustawa uspójniająca pojęcia wykorzystywane w polskim prawodawstwie.

Faktycznie powinny poruszać nas też inne tematy, m.in. sytuacja niektórych spółek Skarbu Państwa czy obszarów strategicznych, gdzie faktycznie kontrola państwowa jest często niezbędna - ale tylko w tych konkretnych obszarach. Górnictwo, jeden z najważniejszych obszarów.

Jedziemy dalej. Te składy jeżdżą do dzisiaj, bez modernizacji. Pisałem do ówczesnego prezesa spółki Przewozy Regionalne, pytałem, co z modernizacjami. Dostałem mało konkretną odpowiedź, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Czyli faktycznie jest super. Ciekawe, czy coś się tutaj zmieni, bo pieniądze na to będą. I rzecz najbliższa mojemu sercu, czyli przemysł stoczniowy, jeśli w ogóle możemy o takowym jeszcze w Polsce mówić. To, co zrobiliście z ludźmi pracującymi m.in. w Gryfii w Świnoujściu, woła po prosu o pomstę do nieba. 200 osób dostało zwolnienia, tym samym ludzie kooperujący z tą stocznią, łącznie ok. 1 tys. osób, w zasadzie stracą pracę, i to w sytuacji, kiedy stocznia była po prostu rentowna. To jest analfabetyzm ekonomiczny. Takie rzeczy może zrobić politolog, ale nie powinno tak się dziać na stanowiskach kierowniczych właśnie w zakładach spółek Skarbu Państwa. Teraz druga stocznia, bliższa mi, bo z naszej okolicy, z Trójmiasta, stocznia Nauta. Stocznia jest w restrukturyzacji, nie wiadomo, co z tym zrobić, długi nie są spłacane. To są sprawy, którymi należy się zająć. Jeśli będziecie na najważniejsze stanowiska wpuszczać kolegów kolegów i koleżanki koleżanek, to w Polsce nigdy nie będzie lepiej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Artur Dziambor ze zjedzonym przez swojego przyjaciela z koła czasem. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Patrzymy na to, co się dzieje, i troszkę nas mrozi. Wczoraj Konfederacja zorganizowała konferencję prasową w sprawie stoczni w Świnoujściu.

Trzeba było to zwyczajnie sprzedać, nie zamykać, ponieważ macie taką fanaberię, bo jeden z waszych byłych posłów, który został tam prezesem, po prostu spieprzył robotę. Trzeba było to sprzedać na prywatnym rynku, podobnie jak większość spółek Skarbu Państwa. Wystarczy nie kraść, bo tak się obsadziliście w tych spółkach Skarbu Państwa, powrzucaliście tam przyjaciół, rodziny, wszystkim jest tam dobrze, ciepełko tam mają, mają wysokie stanowiska z wysokimi wypłatami. To są te synekury, których powinniście się pozbyć. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Rozpoczynamy. Tak, dziękuję bardzo. Oczywiście te zmiany powinny być dokonane, natomiast mam pytanie do ministerstwa, czy nie czuje się źle z tą całą sytuacją, ponieważ mamy sytuację absurdalną. Mamy sytuację polegającą na tym, że są nie drobne zmiany, ale zwyczajnie błędy w dwóch ustawach.

Dziękuję.

Pan poseł Mieczysław Kasprzak z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Odnoszę takie wrażenie, że pani posłanka Kretkowska zapomniała zadać pytanie, ale czas poleciał. Obywatele mówią nam, co mamy poprawić w prawie, a moje pytanie brzmi: Czy rząd przeprowadza takie analizy?

Czy rząd coś takiego robi? A drugie pytanie brzmi: Jaka jest dzisiaj faktyczna sytuacja LOT-u? Bo z tego, co wiemy, to ona jest dramatyczna. Co dalej z LOT-em? Bo akurat ta ustawa dotyczy Polskich Linii Lotniczych LOT. Co dalej z LOT-em? Praktycznie wszystko zamarło. Jaka jest dzisiaj sytuacja, panie ministrze, jeżeli chodzi o LOT? Dziękuję serdecznie. Pani poseł Joanna Fabisiak. Nie ma pani poseł? Zapraszam serdecznie. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Mamy armię urzędników w ministerstwach, którzy nie wychwycili błędów w ustawie, zrobił to obywatel, za co należą mu się słowa uznania i podziękowania.

Wnieśliśmy w tej sprawie poprawkę. A propos powołań i odwołań. Szanowni państwo, od wczoraj w Porcie Lotniczym Lublin pracuje, została powołana do rady nadzorczej szwagierka wiceministra Sasina. Mam pytanie do pana ministra. Czy powołanie szwagierki będzie się wiązać z tym, że Port Lotniczy Lublin dostanie pomoc i wsparcie w ramach tarczy 2.0, ponieważ zostało to usunięte z tej tarczy? Mam nadzieję, że obecność tej pani przysłuży się lotnisku, a nie będzie tylko kosztem. Dziękuję. Ciekawe pytanie. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Konrad Berkowicz, koło Konfederacji. Zapraszam, panie pośle. Na wstępie przepraszam wyborców, że występuję zamaskowany, ale to nie dlatego, że dołączam do sejmowych bandytów, tylko dlatego, że długo czekałem, aż Prezydium Sejmu się opamięta. Ale niestety ze zdrowym rozsądkiem wygrała wiara w bawełniane maseczki i inne aluminiowe czapeczki i muszę brać udział w przymusowym balu maskowym, mimo że mówię raptem do ośmiu posłów na sali, którzy są w odległości kilkudziesięciu metrów ode mnie. Natomiast mówimy o państwowych przedsiębiorstwach, które różnią się od prywatnych przedsiębiorstw tym, że nie mogą zbankrutować, bo opierają się na budżecie państwa, na podatkach obywateli. Nie kierują się rachunkiem zysków i strat, bo nikt na tym nie zarabia - albo państwo traci, albo nie traci, jak traci to po prostu zwiększa podatki. W związku z tym pytanie do pana ministra: Czy nie uważa pan, że państwowe przedsiębiorstwa należałoby oddać prywatnym właścicielom tak, żeby nie marnować pracy ludzi ciężko pracujących (Dzwonek) w tych przedsiębiorstwach i żeby całe społeczeństwo zyskało? Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Wie pan, muszę skomentować pana słowa.

moim bardzo bliskim znajomym, który o mały włos przez to, że m.in. nie nosił maseczki, nie umarł. I jak pan już się z nim podzieli tą refleksją, to niech pan przemyśli to i zastanowi się, co będzie pan mówił. Zapraszam podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pana ministra Andrzeja Śliwkę. Proszę, panie ministrze. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo! Przedkładany projekt obejmuje wyłącznie zmiany o charakterze porządkującym. Nie mają one charakteru merytorycznego i są oczywistą konsekwencją zmian dokonanych w systemie prawnym na przestrzeni ostatnich lat. Efektem tej nowelizacji jest poprawa spójności, przejrzystości prawa. Jest to wynikiem wniosku obywatela, za co mu serdecznie dziękujemy. Mając na uwadze powyższe, Rada Ministrów pozytywnie opiniuje ten komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy. A odnośnie do pytań informuję pana posła Kasprzyka, że prowadzone są systematycznie analizy związane z przepisami prawa i przy kolejnych nowelizacjach w oczywisty sposób te przepisy są na bieżąco systematyzowane. Co do pozostałych pytań, panie marszałku, jeżeli jest taka możliwość, to odpowiem w formie pisemnej. Jest taka możliwość, panie ministrze. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będą uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. (druki nr 680 i 721) Bardzo proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoki Sejmie! W imieniu Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych przedstawiam sprawozdanie połączonych komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., druki sejmowe nr 680 i 721. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, skierowała 16 października br. powyższy projekt ustawy do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych do pierwszego czytania. Połączone komisje po przeprowadzeniu pierwszego czytania i zapoznaniu się z opinią Biura Analiz Sejmowych oraz po rozpatrzeniu tego projektu ustawy z dnia 29 października 2020 r. uznały, że projekt ten przyspiesza i usprawnia proces rozwiązywania dotychczasowych dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami Unii Europejskiej, co jest niezbędne, gdyż zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na państwach Unii Europejskiej ciąży obowiązek usunięcia tych umów, gdyż sprawy te już rozstrzygają przepisy wewnętrzne Unii Europejskiej, które są często różne od tych traktatów. Już obecnie niektóre ich klauzule arbitrażowe są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Dlatego też połączone Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Spraw Zagranicznych wnoszą, aby Wysoka Izba raczyła uchwalić projekt niniejszej ustawy z druku nr 680 bez poprawek. Dziękuję serdecznie. Zapraszam.

Proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., druki nr 680 i 721. Tak jak powiedział mój przedmówca, na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych połączone komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt, ponieważ jest to projekt porządkujący, projekt, który jest potrzebny wszystkim inwestorom działającym na terenie państw Unii Europejskiej. Projekt ten dotyczy zapewnienia inwestorowi i jego inwestycjom z państwa strony umowy na terytorium państwa drugiej strony umowy ochrony oraz możliwości dochodzenia roszczeń przed międzynarodowym trybunałem inwestycyjnym na podstawie klauzul arbitrażowych inwestor - państwo. Nadmienię, że porozumienie to podpisały 23 państwa europejskie.

Nadmienię również, że połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej umowy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Marta Wcisło, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Zapraszam. Mam przyjemność w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. Jego powstanie związane jest z kwestią traktatów inwestycyjnych zawartych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, tzw. umów intra-EU BIT, które zapewniają inwestorowi i jego inwestycjom z państwa strony umowy na terytorium państwa drugiej strony umowy ochronę oraz możliwość dochodzenia roszczeń przed międzynarodowym trybunałem inwestycyjnym. Szanowni Państwo! Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej porozumienia takie były stosunkowo korzystne.

W zakresie tych umów pojawiały się także wątpliwości. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że wymienione umowy dwustronne bądź pokrywają się z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bądź są z nim sprzeczne. Potwierdzeniem powyższego jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 marca 2018 r., w którym TSUE stwierdził, że klauzule intra-EU BIT są niezgodne z prawem Unii Europejskiej jako naruszające autonomię prawa Unii Europejskiej. Wyrok ten stał się przyczyną tego, że państwa Unii Europejskiej rozpoczęły wypowiadanie umów intra-EU BIT. Polska uczestniczyła w pracach nad ogólnym rozwiązaniem kwestii tych umów. Wynikiem tych prac jest porozumienie, które zostało zawarte 5 maja 2020 r. przez 23 kraje członkowskie. Ponieważ mam 3 minuty, muszę się streszczać. Porozumienie to kończy obowiązywanie umów intra-EU BIT oraz wygasza ich klauzule przedłużonego obowiązywania. Porozumienie stanowi, że klauzule arbitrażowe w sporach między inwestorem a państwem są sprzeczne z traktatami Unii Europejskiej i w związku z tym nie mają zastosowania, nie mogą one stanowić podstawy prawnej do postępowań arbitrażowych. Inwestorowi na zasadach szczegółowo określonych w porozumieniu będzie przysługiwało prawo skierowania sprawy do sądu krajowego, jednakże pod warunkiem, jakim jest wycofanie się inwestora z postępowania arbitrażowego i zrzeczenie się wszelkich praw i roszczeń wynikających z umowy intra-EU BIT. Takie rozwiązanie, szanowni państwo, jest szybsze i tańsze. W uzasadnieniu [[Dzwonek]] projektu ustawy ratyfikującej wskazano, że obecnie polskie sądownictwo jest niezawisłe i niezależne oraz daje inwestorom gwarancję ochrony inwestycji z możliwością dochodzenia swoich praw w Polsce. Bardzo bym chciała, aby tak było. Dziękuję serdecznie, pani poseł. Zapraszam pana posła Andrzeja Szejnę z klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w wyroku wydanym w dniu 6 marca 2018 r. w sprawie Achmea BV przeciwko Republice Słowacji, że klauzule arbitrażowe inwestor - państwo zawarte w umowach intra-EU BIT są niezgodne z prawem UE, gdyż naruszają autonomię prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z tym wyrokiem na państwach członkowskich Unii Europejskiej ciąży obowiązek usunięcia tych umów, łącznie z klauzulami przedłużonego ich obowiązywania, z obrotu prawnego w celu zagwarantowania pewności prawa. Porozumienie ma na celu dostosowanie stanu prawnego do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Achmea. Obowiązywanie tych umów zostało zakwestionowane również przez Komisję Europejską z uwagi na ich niezgodność z prawem Unii Europejskiej. Komisja Europejska wszczęła formalne postępowania w sprawie niezgodności tych umów z prawem przeciwko Austrii, Niderlandom, Słowacji, Szwecji, Rumunii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Natomiast przeciwko pozostałym państwom członkowskim, w tym przeciwko RP, prowadziła nieformalne postępowania, tzw. EU Pilot, i rozważa obecnie wszczęcie formalnych postępowań. W ramach EU Pilot Komisja Europejska zgłasza poważne obawy, że umowy intra-EU BIT jako takie, a także ich poszczególne postanowienia pokrywają się z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub mogą być z nimi sprzeczne. Związanie się porozumieniem nie powinno mieć konsekwencji politycznych. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, które są stronami tych umów, zostały wezwane przez Komisję Europejską do zakończenia obowiązywania tych umów. Porozumienie nie będzie miało negatywnych skutków społecznych i może zostać pozytywnie przyjęte z uwagi na publiczną krytykę w RP umów intra-EU BIT i międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego funkcjonującego na ich podstawie. Zawarcie porozumienia nie powinno wpłynąć na stosunki gospodarcze między RP a pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Umowy intra-EU BIT, których stroną jest RP, zostały zawarte, kiedy Rzeczpospolita Polska nie była członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście pojawia się pytanie, czy niedostateczny dostęp do niezawisłego sądownictwa w RP da inwestorom zagranicznym gwarancję ochrony inwestycji z możliwością dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Takie gwarancje mają polscy inwestorzy na pozostałych rynkach, w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ministerstwo Rozwoju odnotowało tylko trzy przypadki skorzystania przez polskich inwestorów z ochrony przewidzianej tymi umowami przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi. Zawarcie porozumienia w zakresie rozwiązania umów intra-EU BIT czy też klauzul przedłużonego obowiązywania umów już wypowiedzianych nie naruszy polskiego porządku prawnego i doprowadzi do usunięcia niezgodności tych umów i klauzul przedłużonego ich obowiązywania z prawem Unii Europejskiej. Dlatego w imieniu klubu Lewica wnoszę o przyjęcie tego porozumienia i wniosku Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Mieczysława Kasprzaka z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zabierając głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści, chcę powiedzieć, że poprzemy ten projekt, gdyż on wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, jest to korzystne rozwiązanie, robimy krok do przodu. Nie powinniśmy. Zresztą 23 kraje europejskie poparły to rozwiązanie. Ale zmierzam do czego innego.

Jeżeli przedsiębiorcy mają dochodzić swoich praw na rynku naszym, krajowym, na rynku europejskim, a na pewno się zdarzają takie sytuacje, to powinna być uznawalność prawa. To jest właśnie przykład praworządności.

To daje gwarancję, bezpieczeństwo naszym przedsiębiorcom. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Ponieważ widzę, że państwu na tym zależy, to chciałem powiedzieć, że pan poseł reprezentuje Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści. Przyzwyczajamy się do nowej nazwy. Proszę państwa, wchodzimy. Proszę bardzo, wchodzimy w zakres zadawania pytań. Na pytanie jest minuta. Zaczynamy. Proszę bardzo. Nie ma.

Niezwykle ważny projekt ustawy, projekt o ratyfikacji porozumień dwustronnych, ważny dla Polski, ważny dla inwestorów. Ale projekt ważny w kontekście tego, co jest dzisiaj i co będzie w przyszłości, który daje możliwość skrócenia drogi prawnej w przypadku sporów państwo -inwestor. Niestety nie w Polsce. Od dawna wiemy i z różnych stron płyną sygnały, że praworządność w Polsce nie wygląda dobrze. Komisja Europejska, obywatele wydali druzgocącą opinię związaną z tzw. reformą wymiaru sprawiedliwości, która de facto jest deformą. Moje pytanie brzmi: Czy to nie są aby podwójne standardy? Bo obawiam się, że do czasu zakończenia rządów PiS na horyzoncie naszego kraju nie pojawią się inwestorzy, którzy będą (Dzwonek) swobodnie inwestować w naszym kraju, mając na uwadze to, że na czele wymiaru sprawiedliwości stoi polityk. Bardzo dziękuję.

Chcę zadać pytanie, które nie mieściło się w moim wystąpieniu klubowym, mianowicie takie. Obserwując to, co dzieje się dzisiaj, czyli te nieszczęsne negocjacje i zagrożenie wetem, to obniżenie zaufania do Polski jako kraju praworządnego, to obniżenie zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości, cieszę się, że państwo opieracie - i to jest słuszne - zmiany i tekst tego porozumienia na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale dlaczego nie przestrzegacie innych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, chociażby tych, które dotyczą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że dzisiaj inwestorzy zagraniczni, którzy będą oddani w kwestiach spornych i nie będą mieli możliwości przeniesienia tego sporu na poziom arbitrażu międzynarodowego, a tylko na poziom sądownictwa polskiego, będą mieli wątpliwości co do tego, czy inwestować w Polsce i czy w Polsce będą się czuli bezpiecznie? Czy wy zdajecie sobie sprawę, że wszystko, co robicie dzisiaj, co się dzieje na naszych oczach, jest szkodliwe dla inwestycji (Dzwonek) zagranicznych w Polsce? Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Lista posłów zapisanych do pytań wyczerpała się.

Wysoka Izbo! Chciałbym na wstępie stwierdzić, że nie mamy sygnałów świadczących o tym, jakoby inwestorzy zagraniczni mieli ograniczone zaufanie do polskiego sądownictwa i w związku z tym mieli obiekcje co do konieczności kierowania swoich spraw do polskich sądów, to po pierwsze. Po drugie, zwracam uwagę, że to porozumienie służy właśnie temu, aby niezależnie od procedur krajowych można było każdy spór o charakterze inwestycyjnym poddać pod orzecznictwo sądów unijnych, ewentualnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Wysoki Sejmie! W nawiązaniu do omawianego dzisiaj porozumienia należy podkreślić, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał klauzule arbitrażowe wynikające z dwustronnych porozumień pomiędzy poszczególnymi państwami za niezgodne z prawem Unii Europejskiej i to ze skutkiem wstecznym. W przypadku nowych państw członkowskich, a więc i Polski, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skutkuje od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wyrok ten skutkuje w odniesieniu do wszystkich postępowań arbitrażowych inwestor - państwo prowadzonych wcześniej na podstawie umów dwustronnych, czyli umów intra-EU BIT, których obowiązywanie kończy wynikające z ustawy porozumienie.

Czeka nas więc tutaj dosyć duże porządkowanie spraw wynikających z tego porozumienia i w związku z tym to porozumienie jest bardzo ważne, gdyż kończy obowiązywanie dotychczasowych umów dwustronnych bez konieczności - co jest bardzo ważne - ich wypowiadania. Porozumienie uznaje za wygaszone, dlatego też ważna jest jak najszybsza ratyfikacja tego porozumienia. Dlatego też bardzo dziękuję wszystkim posłom i stronie rządowej za sprawne procedowanie nad ustawą. Bardzo dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku (druki nr 688 i 726) Proszę pana posła Artura Łąckiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Słychać mnie, rozumiem? Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 r., druk nr 688.

Celem porozumienia, podobnie jak innych podobnych umów międzynarodowych, było stworzenie ram dla rozwoju i wzmocnienia współpracy handlowej pomiędzy jego sygnatariuszami.

Obecnie nie stosuje się tej metody określenia pojemności statków, jej stosowanie zostało zarzucone 18 lipca 1982 r., tj. w dniu wejścia w życie międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r. Jednakże o ile nie zostanie wymówione po upływie tego terminu, będzie ono przedłużone w drodze milczącej zgody na czas nieograniczony i będzie mogło być wymówione w każdym czasie. W wypadku wymówienia pozostanie w mocy jeszcze przez trzy miesiące od dnia, w którym jedna z Wysokich Układających się Stron zawiadomi drugą o zamiarze uchylenia jego działania” Dziś, bez mała po 100 latach, jako jedna z Wysokich Układających się Stron czynimy kolejny krok do wypowiedzenia tego porozumienia podpisanego w imieniu strony polskiej przez Jego Ekscelencję pana dra Tadeusza Stanisława Grabowskiego, posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego w Sofii. Dla mnie prace nad tą ustawą były okazją do uświadomienia sobie wagi i trwałości prawa stanowionego przez parlament, tego, z jaką rzetelnością i starannością winniśmy my, posłowie, pracować nad podejmowanymi ustawami i jaką odpowiedzialność ponosimy przed historią. Choć nie wiemy, czy wiele ustaw uchwalanych w iście sprinterskim tempie przez Sejm IX kadencji pozostanie ustawami aktualnymi przez prawie 100 lat, czy posłowie 59. kadencji będą mieli okazję którąś. Wysoka Izbo! Wypowiedzenie porozumienia pozwoli na usunięcie z polskiego systemu prawnego aktu prawa międzynarodowego niezgodnego z prawem Unii Europejskiej oraz niestosowanego od dłuższego czasu. Kwestie objęte postanowieniami porozumienia po jego wypowiedzeniu będą regulowane prawem Unii Europejskiej oraz innymi umowami międzynarodowymi, których stronami są Rzeczpospolita Polska oraz Republika Bułgarii. Nie wywoła to negatywnych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych ani politycznych. Z uwagi na kwestie przedstawione powyżej należy uznać wypowiedzenie porozumienia za w pełni uzasadnione. Porozumienie nie realizuje obecnie celu swojego zawarcia, nie jest stosowane w relacjach pomiędzy stronami oraz jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Mając powyższe na uwadze, w imieniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy. Połączone komisje przyjęły rządowy projekt ustawy przez aklamację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Jerzy Materna, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do rządowego projektu ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku, druki nr 688 i 726. Połączone Komisje: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Spraw Zagranicznych rozpatrzyły projekt ustawy w dniu 3 listopada i przyjęły projekt ustawy bez głosu sprzeciwu. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie!

Pozostałe artykuły, które wymieniłem, mają charakter w dużej mierze historyczny i są regulowane innymi aktami prawa międzynarodowego, jak np. prawem Unii Europejskiej czy Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Wypowiedzenie porozumienia nie wywoła negatywnych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych ani politycznych. Jego wypowiedzenie pozwoli na usunięcie z polskiego systemu prawnego aktu prawa międzynarodowego niezgodnego z prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z wspomnianym wcześniej art. 18 porozumienia jego wypowiedzenie możliwe jest w każdej chwili, w każdym czasie. W przypadku wypowiedzenia porozumienia pozostanie ono w mocy przez 3 miesiące od dnia, w którym jedna ze stron umowy zawiadomi drugą o zamiarze wypowiedzenia. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera projekt ustawy i będzie głosować za jego uchwaleniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi pan poseł Arkadiusz Marchewka. Proszę bardzo.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Trzeba przyznać, że jest to dokument, który ma już prawie 100 lat, i kiedy popatrzy się na jego zapisy, na umowę z 1925 r., to znajdzie się tutaj wielkie nazwiska.

Ta umowa międzynarodowa, którą stanowi Porozumienie Prowizoryczne w sprawach handlowych i nawigacyjnych, została podpisana w 1925 r. Oczywiście jej celem było stworzenie ram dla rozwoju i wzmocnienia współpracy handlowej pomiędzy państwami, które tę umowę podpisały. Wprowadzono w niej zasadę tzw. najwyższego uprzywilejowania względem osób fizycznych i prawnych, które pochodzą z państwa strony porozumienia i prowadzą na terytorium drugiego państwa działalność handlową, przemysłową czy też uprawiają żeglugę. Wiele lat później, w 2007 r., doszło do podpisania protokołu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o przeglądzie umów dwustronnych. To porozumienie zachowało swoją moc jedynie w części regulującej kwestie związane z żeglugą handlową, a także rybołówstwem. Pozostałe w mocy przepisy mają w dużej mierze, przede wszystkim charakter historyczny i dziś są regulowane innymi aktami prawa międzynarodowego, zarówno prawem Unii Europejskiej, jak również umowami międzynarodowymi, które dotyczą kwestii morskiej i są zawierane pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Część z tych założeń, część z zapisów tych umów jest dziś niezgodna z prawem Unii Europejskiej, więc wypowiedzenie tej umowy jest w pełni zasadne. Dlatego w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej przedstawiam opinię o poparciu tego projektu ustawy. Wszystkim państwu zainteresowanym historią polecam zapoznanie się z tymi zapisami, bo jest to bardzo ciekawy, prawie 100-letni dokument. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Pan poseł Andrzej Szejna przedstawi stanowisko klubu parlamentarnego Lewica. Wysoka Izbo! Umowa międzynarodowa, jaką jest Porozumienie Prowizoryczne w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, to bez cienia wątpliwości cenny, ale już relikt prawa międzynarodowego i sztuki dyplomacji.

Sejm również ratyfikował konkordat ze Stolicą Apostolską, a oczywiście lewica, czyli Polska Partia Socjalistyczna, głosowała przeciw.

Obowiązujące przepisy porozumienia mają w dużej mierze charakter historyczny, a kwestie w nich zawarte są regulowane innymi aktami prawa międzynarodowego - przez prawo Unii Europejskiej oraz umowy międzynarodowe dotyczące kwestii morskich zawierane w ramach działalności Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Nie zmienia to faktu, że część obowiązujących przepisów jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej, m.in. art. 11 ust. 6 porozumienia dotyczący rybołówstwa. Jak wiemy, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zalicza rybołówstwo do obszarów kompetencji dzielonej między Unią Europejską a państwami członkowskimi, a zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa do obszarów wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej. Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą zatem rezerwować dla siebie uprawnień do korzystania z zasobów rybołówczych, które stanowią własność wspólną. Ponadto wspomniany artykuł narusza ustanowioną w prawie Unii Europejskiej swobodę świadczenia usług w transporcie morskim. Wypowiedzenie porozumienia pozwoli na usunięcie z polskiego systemu prawnego aktu prawa międzynarodowego niezgodnego z prawem Unii Europejskiej oraz niestosowanego od dłuższego czasu. Stan prawny po wypowiedzeniu porozumienia nie ulegnie zmianie, ponieważ, jak już wspominałem, kwestie objęte postanowieniami porozumienia będą regulowane prawem Unii Europejskiej oraz innymi umowami międzynarodowymi, których stronami są Rzeczpospolita Polska oraz Republika Bułgarii. Klub parlamentarnym Lewica oczywiście poprze projekt ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofii dnia 29 kwietnia 1925 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana posła Władysława Teofila Bartoszewskiego o przedstawienie stanowiska Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Słynny angielski minister spraw zagranicznych i premier lord Palmerston powiedział kiedyś: Wielka Brytania nie ma wiecznych wrogów i niezmiennych przyjaciół, ma natomiast wieczne i niezmienne interesy i za tymi interesami będziemy podążać. Polska nie była tak szczęśliwa jak Wielka Brytania, bo przez 200 lat historii nie mieliśmy samodzielnej polityki zagranicznej w związku z okresem zaborów, z okresem II wojny światowej i dominacji sowieckiej przez kilkadziesiąt lat w Polsce. Mieliśmy tylko 20 lat szczęśliwych, kiedy to nasza polityka zagraniczna była suwerenna. Z wielką przyjemnością dowiedziałem się, że obowiązuje nas do tej pory Porozumienie Prowizoryczne w sprawach handlowych podpisane, zawarte pomiędzy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a królem Bułgarów. Jest to unikalny dokument, ponieważ ma prawie 100-letnią już historię. Jest rzeczą jak na polskie warunki niesłychaną, że obowiązuje nas sześć artykułów tego porozumienia, które do tej pory jest ważne. To jest przyczynek do historii dyplomacji polskiej bardzo interesujący. Z wielkim wzruszeniem zobaczyłem, że ten dokument został ratyfikowany przez prezydenta Mościckiego, premiera Piłsudskiego i ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego. Jest rzeczą oczywistą, że Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska przychyla się do tego, żeby to Porozumienie Prowizoryczne wypowiedzieć, bo jest to dokument o charakterze w tej chwili czysto historycznym i w związku z tym nie powinien dalej obowiązywać. Jest on sprzeczny z prawem unijnym. Szczerze mówiąc, żaden poseł z żadnego ugrupowania nie wniósł jakichkolwiek obiekcji ani nie zadał pytań co do tego. Zakładam, że tak będzie teraz na sali sejmowej. Dziękuję bardzo panu posłowi. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Robert Winnicki. Wysoka Izbo! Trzy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w przypadku tego dokumentu. Pierwsza to uwaga historyczna. Oczywiście pan poseł Bartoszewski ma rację, mówiąc o tym, kto ratyfikował, ale kto negocjował ten traktat, to porozumienie? Przede wszystkim rząd Władysława Grabskiego, jednak wcześniejszy rząd, w tym m.in. przez 7 miesięcy urzędujący na funkcji ministra spraw zagranicznych hrabia Maurycy Zamoyski. Czyli politycy Narodowej Demokracji ten dokument negocjowali.

Warto na ten aspekt historyczny zwrócić uwagę, szanowni państwo, dlatego że polskie biuro prasowe w Bułgarii zaczęło działać już w 1915 r., 3 lata przed odzyskaniem niepodległości, 4 lata tak naprawdę przed uformowaniem się dyplomacji polskiej w jej skrystalizowanej formie, 4 lata przed kongresem w Wersalu. Ten kierunek bałkański nie był zaniedbywany w tamtym okresie, i bardzo dobrze, a ta przenikliwa działalność wybitnego profesora i dyplomaty jest tutaj szczególnie nie do pominięcia. Szanowni Państwo!

Ale nie wolno zaniedbywać tego regionu, w którym możemy realizować swoje interesy i mamy dużą życzliwość i dużo przyjaciół, którzy potencjalnie mogą z nami współpracować. Tutaj widzę dużo do nadrobienia, jeśli chodzi o polską dyplomację. Szanowni państwo, ta umowa, dzisiaj już przechodząca do historii po blisko 100 latach - ale i świeższe przykłady, jak przykład Wielkiej Brytanii - pokazuje nam, jak bardzo ważne jest, żeby suwerenne państwo nie zaniedbywało posiadania kadr dyplomatycznych zdolnych do negocjowania umów gospodarczych, wysoko kompetentnych kadr, które będą w stanie o interesy gospodarcze państwa dbać na arenie międzynarodowej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo panu posłowi. Jeżeli nie ma więcej zgłoszeń, to zamykam listę. Ustalam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Proszę pana posła Mirosława Suchonia o zadanie pytania. Nieobecny. Zatem pan poseł Andrzej Szejna, Lewica. Wysoka Izbo! Oczywiście wspomniałem o ratyfikowaniu konkordatu ze Stolicą Apostolską przy sprzeciwie lewicy w 1925 r. Przypomnę również, że wtedy miał też miejsce upadek rządu pana premiera Grabskiego. Później był pan premier Skrzyński, a potem był pan premier Witos. Oczywiście to też są bardzo ważne w historii Rzeczypospolitej Polskiej lata, które później pokazały, że jednak miejsce Polski jest w Europie. Broniliśmy również w pewnym sensie Europy przed nawałą sowiecką, broniliśmy naszego miejsca, naszych korzeni, naszej historii, naszej świeżej niepodległości. Moje pytanie jest takie: Czy właśnie z tych historycznych wydarzeń, które nastąpiły już później, nie wyciągacie państwo wniosków co do swojej dzisiejszej polityki, która polega na izolacji Polski w Europie, na odosobnieniu? I drugie pytanie: Dlaczego (Dzwonek) tak długo czekaliśmy na dostosowanie prawa polskiego i tej umowy do prawa europejskiego? Dziękuję. Bardzo dziękuję.

W związku z tym nie widzę też powodu, aby szerzej rozwijać ten temat. Mamy bardzo ścisłą współpracę z wieloma krajami europejskimi i pozaeuropejskimi. Transatlantyckie relacje też są bardzo dobre. Natomiast dlaczego tak długo czekaliśmy na ratyfikację?

Ten projekt, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest częścią właśnie tego programu.

Proszę teraz pana Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, o odniesienie się, jeżeli jest taka potrzeba. Też wiemy, że nie. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 808) Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, głównego geologa kraju, pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej państwa pana Dziadzia o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

Szanowni Państwo! Panie Marszałku! Chciałbym przedstawić państwu projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który stanowi zwieńczenie kilkuletnich prac nad inteligentnym opomiarowaniem w energetyce oraz usprawnieniem funkcjonowania krajowych rynków energetycznych. Szanowni Państwo! Ustawa stanowi niezbędny punkt wyjścia do transformacji sektora energetycznego opartej m.in. na jego cyfryzacji, inteligentnych sieciach, inteligentnych licznikach zdalnego odczytu. Ustawa umożliwi bezpieczną integrację odnawialnych źródeł energii w systemie oraz wykorzystanie energii w sektorze, w tym zwiększenie elastyczności systemu energetycznego, a także wykorzystanie potencjału aktywnych odbiorców. Celem projektu jest zapewnienie ram dla funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania w energetyce poprzez zainstalowanie do 2028 r. inteligentnych liczników u co najmniej 80% odbiorców, powołanie operatora informacji rynku energii odpowiedzialnego za prowadzenie systemu zbierającego i przetwarzającego informacje i dane pomiarowe z tych zainstalowanych liczników, tzw. centralnego systemu informacji rynku energii.

Projekt zawiera również kompleksowe rozwiązania w zakresie usuwania bariery prawnej dla rozwoju magazynów energii umożliwiające dalszy rozwój energetyki rozproszonej, tzw. energetyki prosumenkiej, i OZE, zwiększenia ochrony konsumentów na rynku energii i paliw gazowych m.in. przez zakaz zawierania umów za pośrednictwem sprzedawców energii i gazów w formie akwizycyjnej, tzw. door-to-door, ułatwień dla działalności przedsiębiorstw energetycznych, m.in. wprowadzenia instytucji zamkniętych systemów dystrybucyjnych i rozwiązań dla pojazdów trakcyjnych, oraz usprawnienia kontroli nadzoru nad rynkiem energii, paliw gazowych, paliw ciekłych przez szerokie wzmocnienie nadzoru URE. Przyjęcie tej ustawy przez Sejm będzie milowym krokiem dla rozwoju polskiej energetyki przyszłości. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Przystępujemy teraz do przedstawienia stanowisk klubów parlamentarnych i koła. Jako pierwszy zabierze głos pan poseł Witold Czarnecki i przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że zmiany obejmują 20 obszarów objętych dotychczasowym działaniem ustawy. Omówiony projekt ustawy dostosowuje przepisy polskiego prawa do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

Ponadto według tego projektu ustawy to prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących pracę przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych. Z ustawą wprowadza się przepisy, na podstawie których prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł cofnąć koncesję w przypadku wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorcy energetycznego decyzji o uznaniu praktyki działań tegoż przedsiębiorstwa za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Projekt ustawy prowadzi do urealnienia kosztów ponoszonych przez właścicieli pojazdów oddających energię elektryczną do sieci trakcyjnej w następstwie ich hamowania, co odzwierciedla rzeczywiste zużycie energii. Projekt ustawy wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii, usprawnia też funkcjonowanie systemów inteligentnego opomiarowania, o czym mówił pan minister, w sieci elektrycznej dzięki wprowadzeniu rozliczeń gospodarstw domowych tak, by były one rozliczane za energię elektryczną rzeczywiście zużytą, a nie prognozowaną. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i rekomenduje skierowanie do dalszych prac w wersji, która została paniom i panom posłom wręczona w druku sejmowym nr 808. Dziękuję bardzo panu posłowi. Pan poseł Tomasz Piotr Nowak przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! To była bardzo ciężka noc. Wczoraj o godz. 21 dowiedzieliśmy się, że mamy przestudiować 1429 stron po to, ażebyśmy dzisiaj mogli przedłożyć sprawozdanie. Nad tego typu ustawami pracuje się co najmniej pół roku w parlamentach, które szanują proces legislacyjny. Ustawa była zakończona, konsultacje były zakończone w lipcu 2018 r. i nie rozumiem, dlaczego półtora roku czekało się na to, ażeby ustawa trafiła do Sejmu i żeby nad nią tutaj obradowano.

Na Prawo energetyczne czekamy od dawna. Nie ma przeniesienia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostaw na OSD i np. na lokalne rynki czy lokalne bilansowanie. Nie ma prosumenta zbiorowego i wirtualnego. Na to wszystko czekamy. Mam nadzieję, że pojawi się to za chwilę. Kontrowersje, jakie budzi ta ustawa, to wymogi dużych zabezpieczeń dla spółek obrotu hamujących rozwój konkurencyjny pojawiania się kolejnych spółek obrotu, bowiem blokada będzie ubezpieczeniowa. Centralny system przetwarzania danych przez operatora informacji rynku energii jest kontrowersyjny - o tym za chwilę. Ciekawa jest definicja np. instalacji hybrydowej OZE, która startować będzie w aukcjach w swojej kategorii, ale magazyny energii w ramach tej definicji powinny być własnością tych, którzy startują, a przecież mogłyby być zakontraktowane. To są drobiazgi, ale bardzo istotne. I takich drobiazgów może być wiele, wiele, wiele.

To jest uregulowanie kompleksowe i my się z tym kierunkowo zgadzamy.

Przetwarzanie danych będzie leżało w gestii operatora informacji rynku energii z PSE. Systemy tego typu są scentralizowane lub zdecentralizowane.

Tymczasem tu agregacja danych będzie ogromna i będzie w jednym ręku. Tym bardziej dziwi właśnie w tym momencie fakt, że ustawa nie była konsultowana z prezesem urzędu danych osobowych. Przecież na podstawie zagregowanych danych będzie można stworzyć mapę naszych zachowań, rytmu dnia itd. Jak te dane będą zabezpieczone? Dlaczego prezes urzędu nie zajął tu stanowiska?

Co z biedniejszymi odbiorcami, którzy nie będą sobie mogli pozwolić na ten licznik? Chodzi o to, ażeby przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu, bo ten, kto nie będzie miał tego licznika, siłą rzeczy będzie miał droższą energię.

To jest niezbędne, żeby zrealizować zasadnicze cele tej ustawy, a mianowicie zmniejszyć obciążenie szczytowe, tak żebyśmy konsumowali tę energię nie w szczycie, tylko w innych przedziałach czasu, aby ten szczyt zmniejszyć. Oczywiście my kierunkowo jesteśmy za tą ustawą i chętnie będziemy nad nią pracować. Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana posła Dariusza Wieczorka, aby przedstawił stanowisko klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ale oczywiście nie ma na co narzekać i się skarżyć, bo energetyka to jest jądro polskiej gospodarki i bez energetyki nikt z nas nie może funkcjonować.

Oczywiście pojawia się kilka dobrych zapisów dotyczących rzeczywiście pójścia wreszcie w nowe technologie, a więc chodzi o kwestię uruchomienia magazynów energii, kwestie dotyczące opomiarowania stacji średniego napięcia i kwestie dotyczące oczywiście opomiarowania odbiorców. Rodzi się tylko pytanie, czy od początku do końca zostało to wszystko wyliczone. Bo prawda jest taka, że jeżeli chodzi o cały ten proces, to wszystkie opracowania, które od 2012 r. są realizowane, mówią o koszcie na poziomie 10 mld zł. Jeżeli mówimy o dzisiejszych czasach i o tych kosztach, które są większe, to pewnie to są również większe koszty.

Jest również pytanie o ustalenie, w jaki sposób te informacje będą wykorzystywane, w jaki sposób one będą wykorzystywane dla dobra rynku energii, bo to jest najistotniejsza sprawa. Już dzisiaj koncerny energetyczne wprowadziły w niektórych miejscach takie pilotażowe rozwiązania, kilkadziesiąt tysięcy tego typu liczników jest założonych. Jest takie pytanie: Czy ta ustawa uwzględnia te doświadczenia? Bo mówimy tutaj nie tylko o samym liczniku, który ma jakąś funkcjonalność, ale mówimy również o całym systemie informatycznym, który będzie obsługiwał te wszystkie informacje. Powstaje pytanie: Czy rzeczywiście te środki, które już zostały wydane, nie zostały wyrzucone w błoto? Czy ta ustawa pozwoli na to, żeby te nakłady również wykorzystać?

Jest pytanie: Jak i kiedy można to stworzyć, jakie będą tego koszty? Bo to znowu będzie musiało się pojawić pewnie w taryfie przedsiębiorstw dystrybucyjnych czy przedsiębiorstwa przesyłowego.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz głos zabierze pan poseł Mieczysław Kasprzak, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści. Panie Marszałku! Zabierając głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści - długa nazwa, ale tak jak mówiłem wcześniej, ona będzie jeszcze dłuższa - chciałbym powiedzieć i potwierdzić, że rzeczywiście jest to ustawa z grupy ustaw ciężkich, może nie dlatego, że jest obszerna, ale problematyka jest ważna, trudna, skomplikowana, wymagająca wielu rozwiązań, które niosą tę innowacyjność. Należy się cieszyć - bo niektórzy narzekają, że ustawa wpłynęła dopiero wczoraj wieczorem - że ustawa wpłynęła, bo mogłaby nie wpłynąć. Znając zachowanie w zakresie energetyki, przez wiele lat obserwujemy, że dobre rozwiązania są blokowane. Mówiąc o energetyce, cały czas mamy na myśli przechodzenie na nowoczesne źródła energii, energii zielonej, energii odnawialnej, energii przyszłości. O tym Polskie Stronnictwo Ludowe od wielu lat mówi i domagamy się tutaj dobrych rozwiązań. Niestety mamy opóźnienia w tym zakresie. Ta ustawa jest oczekiwaną ustawą, bo rozwiązania w zakresie inteligentnego opomiarowania, tego, które powinno być już wprowadzane, są potrzebne. To daje możliwości oszczędzania energii, bo my przez oszczędność energii możemy też - i taki jest cel - ograniczyć emisję, szanować środowisko, szanować atmosferę. Ale to musi być jasne, przejrzyste. Chyba nikt z Polaków nie odczuwa tego, że państwo idzie w kierunku oszczędzania energii przez obywateli. Ten system rozliczeniowy, który mamy w tej chwili, i dostępność tych informacji są tak skomplikowane, że nikt nie jest w stanie ocenić, ile energii zużywa. To musi być już jakiś fachowiec, ktoś, kto się w to zagłębi, ale przeciętny Polak nie jest w stanie sobie tego wyliczyć. Nie ma takich mechanizmów, żeby w danym momencie albo wyłączyć urządzenie, albo zwiększyć zużycie energii. Nie ma systemu, który by pokazywał Polakowi, jak oszczędzać na energii, nawet na cenie energii, bo ta energia może być w różnych godzinach, w różnym czasie dobowym różnie wyceniana.

Ale to nie może być tak jak w tej chwili też w licznikach, że jest kilkadziesiąt danych. I teraz konia z rzędem temu, kto jest w stanie to wszystko przeanalizować. Dzisiaj, w dobie smartfonów, gdy mamy szereg możliwości dostępu do różnej wiedzy, sterowania urządzeniami w różnych miejscach, nie mamy możliwości odczytania tego, co się dzieje w naszym domu w zakresie energii elektrycznej. To powinno być dostępne i w tym kierunku powinniśmy iść, żeby w każdej chwili obywatel mógł widzieć, jak sterować swoimi urządzeniami. Nowoczesne technologie, jeżeli chodzi o gromadzenie energii, to też jest ogromny postęp w tym zakresie. Powinniśmy w tym kierunku zmierzać, aby wchodzić w te nowoczesne technologie i nie bać się tego. Bo często boimy się tego, świat nam ucieka.

Ale dzisiaj już przy tych zmianach, które wchodzą, szczególnie młode pokolenia, myślę, że oczekują na to, aby w zakresie klimatu, w zakresie oszczędzania energii mieć tę możliwość bezpośredniego wpływu, bo to jest bezpośredni wpływ obywatela na to, co może zrobić w zakresie energii elektrycznej. Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści, a szerzej mówiąc: Koalicja Polska będzie chciała aktywnie pracować w tym zakresie, bo to są ważne rozwiązania, ważne propozycje, oczekiwane przez system energetyczny, ale i przez Polaków. Bardzo dziękuję panu posłowi. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Robert Winnicki. Wysoka Izbo! Przedstawiona regulacja oczywiście ma swoje zalety, w wielu obszarach upraszcza zasadę dostępu, upraszcza zasady, na jakich będzie się odbywał chociażby odczyt bez obecności fizycznej inkasenta, upraszcza sprawę odbiorców, którzy będą rozliczani z energii elektrycznej zgodnie z rzeczywistym zużyciem, a nie według prognoz. Rzeczywiście sposób procedowania nad nią jest jak zwykle fatalny. Jutro na szczycie unijnym jednym z tematów będzie po raz kolejny walka z ociepleniem klimatycznym. Szanowni Państwo! Już obecne regulacje, obecnie przyjęte, obecna kapitulacja na poziomie 40% jest bardzo groźnym zjawiskiem dla polskiej gospodarki. Uderza bezpośrednio w naszą energetykę, uderza w nasz przemysł energochłonny. To są propozycje, które nigdy nie powinny być przez Polskę zaakceptowane. Europejski Zielony Ład jest uderzeniem w samo jądro polskiej energetyki i polskiego przemysłu energochłonnego. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. W naszych warunkach energetycznych jest po prostu utopią. Jest to szkodliwa utopia forsowana przede wszystkim przez lobby francuskie i niemieckie. I nie ma innej drogi wyjścia z tej matni, która ma być jeszcze zaostrzana przez brukselskich decydentów i komisarzy, niż wyłączenie się z unijnej, a de facto brukselskiej, berlińskiej, brukselsko-berlińskiej polityki klimatycznej. Nie ma innej drogi. Trzeba po prostu postawić weto, ponieważ to nam zniszczy nasz przemysł i naszą energetykę.

Punkt pierwszy. Punkt drugi. Szybka budowa energetyki jądrowej.

Znaczy, państwo cały czas rozmawiają, państwo cały czas tokują, deliberują. Minęło 5 lat, takie są fakty.

Co więcej, co gorzej, najbardziej zaawansowane rozmowy są ze Stanami Zjednoczonymi. My nie powinniśmy opierać naszej współpracy w zakresie energetyki jądrowej z żadnym dużym mocarstwem mającym różne interesy w różnych częściach świata. My powinniśmy dyskutować z Koreą Południową, dyskutować z Francją, która nie jest supermocarstwem o takich interesach i takich wpływach jak chociażby Stany Zjednoczone. Nie możemy się uzależniać. Nie możemy, uniezależniając się gazowo od Federacji Rosyjskiej, co jest słuszne. Należy zdywersyfikować dostawy gazu z kierunku północnego, z Norwegii, ze Stanów, z Rosji, z Zatoki Perskiej. Tak, to powinno być zdywersyfikowane i ku temu idziemy, Bogu dzięki. Ale nie można w energetyce jądrowej teraz na inne supermocarstwo przekładać wajchy i uzależniać się tak głęboko w zależności już będącej militarną, już mamy zależność militarną bardzo pogłębioną. Przecież to są absurdalne rzeczy, absurdalne kwoty. Nie tylko UE dąży do podnoszenia cen prądu. Od 1 stycznia w życie wchodzi opłata mocowa, co oznacza wyższy comiesięczny rachunek za prąd dla każdego gospodarstwa domowego o ok. 10%. Czy Polacy sobie z tego zdają sprawę? My jako Konfederacja żądamy jasnej, stanowczej polityki energetycznej państwa, planu polityki energetycznej państwa opartego o te (Dzwonek) trzy filary: po pierwsze, stopniowe zmniejszanie udziału węgla, ale racjonalne, po drugie, racjonalne też, zwiększanie udziału energetyki odnawialnej, po trzecie, radykalne i szybkie przejście do sensownego programu jądrowego i przede wszystkim do wypowiedzenia pakietu klimatycznego Unii Europejskiej, ponieważ z nim nasza energetyka, nasz przemysł energochłonny daleko nie zajedzie. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Czy ktoś jeszcze chciałby dopisać się do listy?

Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Anita Sowińska, Lewica. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie pośle Winnicki, szkodliwy to jest pan i denialiści klimatyczni, i płaskoziemcy, to jest tyle. To jest długo oczekiwana ustawa, która zmienia całkowicie system energetyczny. i umożliwia oparcie systemu na odnawialnych źródłach energii. To one, jeżeli będzie wprowadzony dobrze przemyślany system dynamicznych cen energii, umożliwią to, że będziemy mogli magazynować energię wtedy, kiedy będzie jej za dużo, będziemy mogli magazynować energię wtedy, kiedy jest bardzo tania. I w związku z tym mam pytania do pana ministra. Pan minister powiedział, że planuje wymienić 80% liczników do 2026 r., jeżeli dobrze zrozumiałam.

I jakie są źródła finansowania, czy te koszty poniosą operatorzy, czy będą środki z Unii Europejskiej, czy środki z budżetu państwa również w tym są? I jeszcze moje ostatnie pytanie: Jaki jest tryb wyboru prezesa URE? Dziękuję bardzo. Pani chyba nie rozumie rzeczywistości. Sytuacja jest taka, mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi, z których na pewno część jest również pochodną działań człowieka. Cała Unia Europejska, cała Europa to jest 10% w skali światowej. Największe wzrosty, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, nie są w Europie, tutaj mamy raczej stabilność albo redukcję, największe wzrosty są w państwach rozwijających się. Choćby cała Unia Europejska do zera zlikwidowała emisję dwutlenku węgla, co oczywiście jest utopią, nie zmieni to w ogóle sytuacji, jeśli chodzi o klimat na świecie. Jedynym systemowym rozwiązaniem dla klimatu na świecie jest masowe upowszechnienie się technologii jądrowych.

Tak, dziękuję.

Chciałabym przyłączyć się do uwag i zapytań złożonych przez fundację ClientEarth do tej ustawy i zapytać, dlaczego ustawodawca w sposób jedynie wybiórczy powołuje się w uzasadnieniu na nowy pakiet energetyczny. Czy pani poseł, możemy prosić o. Proszę bardzo. Czy ja mogę. Mam zacząć jeszcze raz czy. Proszę kontynuować. Dlaczego ustawodawca w sposób jedynie wybiórczy powołuje się w uzasadnieniu na nowy pakiet prawa energetycznego Unii Europejskiej, tzw. pakiet zimowy, to tzw. czysta energia dla wszystkich Europejczyków, idąc w zasadzie wbrew głównym trendom w tym pakiecie zmian, a te główne trendy to jest umiejscowienie konsumenta w centrum rynku energii i przechodzenie na zeroemisyjny system energetyczny?

Dlaczego zatem nie uwzględnia się zmian przepisów dotyczących taryfowania w tym projekcie, tak aby umożliwić wprowadzenie mechanizmów zarządzania popytem przez odbiorców energii? Dlaczego nie ma wyraźnego wskazania, że politykę energetyczną prowadzi się na rzecz i w interesie właśnie tego odbiorcy energii, czyli konsumenta?

Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Pytanie teraz zada pan poseł Mieczysław Kasprzak, Koalicja Polska. Zabierając głos w imieniu Koalicji Polskiej, chciałem złożyć tutaj pewną deklarację. My jednak będziemy za energią zieloną, energią odnawialną. Mówimy tutaj o wielkich sprawach, o nowoczesnych technologiach, ale dzisiaj problem jest gdzie indziej. Problem jest w sieciach energetycznych. Dzisiaj wiele sieci energetycznych nie jest już w stanie przesyłać prądu, blokuje się. W związku z tym, że wielu prosumentów zainstalowało własne urządzenia fotowoltaiczne na swoich dachach, dzisiaj sieci się blokują. A więc moje pytanie: Czy te 40-, 50-letnie sieci będą remontowane? Jakie środki finansowe Skarb Państwa, spółki skarbu państwa przeznaczą na remont sieci energetycznych? Gdzie są one remontowane (Dzwonek), które spółki remontują, wprowadzają modernizacje sieci energetycznych? Czy będzie procedowany projekt, który oczekuje już od dłuższego czasu na rozpatrzenie, jeżeli chodzi o rynek mocy? Koalicja Polska złożyła wniosek, żeby o rok przełożyć wejście tej ustawy, jeżeli chodzi o opłaty, bo dzisiaj, w dobie pandemii, nie możemy podnosić ceny energii elektrycznej o 15%. Czy ten projekt będzie procedowany w najbliższym czasie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Obiecuję, że o to zapytam na najbliższym posiedzeniu Prezydium Sejmu. A do kolegów posłów miałbym prośbę, żeby jak zadaje pytanie jeden z naszych kolegów, po prostu troszkę wyciszyć te rozmowy. Proszę teraz pana posła Dariusza Kurzawę. Chyba że zdalnie. Nie. W takim razie pytanie zada pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska. I wszyscy będziemy z uwagą słuchali pytania, które zadaje pan poseł. Panie Ministrze! Rzeczywiście oczekiwana ustawa w wielu zapisach jest trochę trudna i kontrowersyjna, natomiast wiele obowiązków w ramach tej ustawy, tych działań, które państwo przedstawiacie, spoczywa na URE, na prezesie URE. Chciałbym zapytać: Czy państwo konsultowaliście, jaka jest opinia prezesa URE dotycząca jego zadań zapisanych w tym projekcie ustawy i ile środków trzeba przeznaczyć dla tego urzędu, żeby cała machina związana z realizacją tej ustawy zadziałała skutecznie? Przecież centralny system przetwarzania danych to jest potężna machina, która będzie zbierała dane właściwie wszystkich, którzy w tym systemie będą uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Mirosława Suchonia. Nie ma. To teraz pan poseł Tomasz Piotr Nowak zada pytanie. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ale proszę powiedzieć: Czy wszystkie uwagi tych podmiotów zostały uwzględnione, a jeśli nie, to jak wyglądał protokół rozbieżności?

Następna sprawa. Jaką wiedzę ma ministerstwo na temat oszustw, które były dokonywane poprzez podpisywanie umów ze spółkami obrotu, które podszywały się pod spółki powszechnie znane, typu Energa, Enea itd.

Bowiem one były prognozowane i później wielu ludzi stawało przed taką sytuacją, że nagle przychodził rachunek wyrównujący i on dotyczył nieraz kilku tysięcy złotych, a kiedy człowiek - miałem takie przypadki i do mnie docierali ludzie z interwencją - zwracał się do spółki operatora, to był odsyłany na tzw. drzewo, czyli nie wytłumaczono mu, na czym polegało to, że nagle zużył tyle energii. Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana posła Wojciecha Saługę o zadanie pytania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To oczekiwana zmiana Prawa energetycznego, bardzo obszerna, wiele spraw poruszanych. Ale też musimy sobie powiedzieć, w jakim otoczeniu ona się dzieje - mamy jedną z wyższych stawek za prąd w Europie, przedsiębiorstwa energochłonne nie wyrabiają po prostu z tą ceną prądu i gaszą produkcję, mamy import węgla z zagranicy, sieci energetyczne nie są w stanie przesyłać prądu, który produkujemy, mamy import energii także rekordowy, a na koniec zamykane jest górnictwo z powodu nieopłacalności produkcji, ale też nieopłacalności produkcji prądu z węgla.

Czy to jest prawo i po prostu te przyłącza będą już legalne od tego czasu, będą legalnie (Dzwonek) działały, czy też w sądach będzie można dochodzić, gdy ktoś się nie będzie z tym zgadzał? Bo samą ustawą nie spowodujemy, że urządzenie pomiarowe będzie działać sprawnie i będzie pokazywać prawdziwe wyniki. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze!

To bardzo dobrze. Wiadomo, że inteligentne liczniki są korzystne dla wszystkich, bo umożliwiają bardziej racjonalne gospodarowanie energią. Są też oczywiście wygodniejsze dla klientów. Unijne uregulowania pojawiły się w systemie prawnym w roku 2012.

W tym czasie spółki energetyczne przestały przynosić zyski. W tym czasie energię mamy chyba najdroższą w Europie. Przy okazji: tak - dla Unii Europejskiej, nie - dla weta. Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana posła Stanisława Żuka, posła niezrzeszonego, o zadanie pytania.

Wysoka Izbo! Może na początku pytanie, bo czasu jest niewiele. Panie ministrze, kiedy rząd przedstawi nową politykę energetyczną Polski?

Dlaczego opowiadacie takie bzdury, że Polska ma najdroższą energię?

Ostatnie zdanie.

Pytanie: Kiedy będzie polityka? Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz pana posła Dariusza Wieczorka o zadanie pytania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozmawiamy o wielkim przedsięwzięciu dla energetyki, czyli o wprowadzeniu inteligentnych liczników.

Czy projekt ustawy i cały ten proces były konsultowane z polskimi przedsiębiorcami, którzy zajmują się tą branżą? Drugie pytanie. Pojawiają się tam zapisy mówiące o tym, że jeżeli operator przesyłowy zmieni właściciela, to może wypowiedzieć pewne umowy. Pytam wprost: Czy to jest przygotowanie do przejęcia PGNiG przez koncern Orlen? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie zada pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polska znalazła się na 34. miejscu na 36 państw OECD w rankingu konkurencyjności systemów podatkowych. Chodzi o to, jak bardzo system podatkowy jest zagmatwany, jaka jest mnogość podatków, podateczków, opłat, danin, składek, akcyz, itd. To jest wstyd. To jest po prostu jakaś hańba.

Macie moc.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Waldemar Sługocki, Koalicja Obywatelska, zada teraz pytanie. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mianowicie zapowiadacie państwo, i tu chciałbym złożyć gratulacje, elektroniczny system zarządzania konsumpcją energii elektrycznej przez konsumentów.

Chciałem zapytać pana, panie ministrze, o koszty. Czy nie zostaną one przerzucone na konsumentów? Po drugie, mówicie państwo o tym, że pobudzi to rynek producentów tych urządzeń oraz informatyków, którzy znajdą atrakcyjne miejsca na rynku pracy. Ale pytanie jest takie: Co z tymi, którzy dzisiaj odczytują liczniki? W jaki sposób te osoby zostaną zagospodarowane? Dziękuję bardzo panu posłowi. Na zadane wcześniej pytania odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, główny geolog kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa pan minister Piotr Dziadzio.

Szanowni Państwo! Wiele zarzutów, wiele informacji, ale też wiele pozytywnych słów usłyszeliśmy tutaj od państwa. Po pierwsze, jesteśmy zgodni co do tego, że ustawa jest nam potrzebna, żeby zrobić skok cywilizacyjny w elektroenergetyce. Było szereg pytań, które ciężko jest tak na pierwszy rzut oka ułożyć i usystematyzować, bo dotyczyły różnych obszarów. Zacznę przede wszystkim od konsultacji. Ustawa, po pierwsze. Czy mogę kontynuować? Ja już kilkakrotnie prosiłem, panie ministrze. Szanowni Państwo! Ustawa była długo procedowana, to prawda, niemniej jednak przeszła wszystkie możliwe szczeble konsultacji.

Ten długi proces pokazuje, jak złożone problemy są ujęte w ustawie i jak złożone problemy ustawa rozwiązuje. Ten długi okres procedowania pokazał, że ona jest przygotowana do tego, żeby ją wdrożyć, żeby ją wprowadzić.

Oczywiście ona będzie konsultowana, będzie dyskutowana w komisjach. Ambitny czas wprowadzania liczników.

To jest taki kluczowy element.

Tak, oczywiście, była, potwierdzam.

Nie mam w tej chwili danych odnośnie do protokołu rozbieżności, ale generalnie możemy państwu udostępnić ten protokół rozbieżności, to nie jest żaden problem.

To jest bardzo istotny element. Są w stanie to wyprodukować, są w stanie to wprowadzić.

To nie przedsiębiorca, tylko ta ustawa gwarantuje bezpieczeństwo odbiorcy. Było tutaj zarzucane i wielokrotnie przedstawiane przez państwa to, że istnieje pewne zagrożenie, brak zrozumienia dla rozliczania poboru energii elektrycznej.

Oczywiście wszystkie inteligentne rozwiązania, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, z których możemy korzystać już poprzez smartfony, są dla nas dostępne.

Co jeszcze z takich bardzo istotnych kwestii?

Musicie państwo mieć taką świadomość.

To jest bardzo istotne i myślę, że wszyscy państwo sobie z tego zdajecie sprawę.

Jeszcze szukam, czy jeszcze coś z tych uwag. Nie, generalnie były one natury ogólnej.

Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw zawarty w druku nr 808 do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 798 i 810) Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 798. Marszałek Sejmu zgodnie z art. 73 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 3 grudnia tego roku powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu wczorajszym, czyli 8 grudnia, wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalił ten projekt ustawy. Kilka słów dodatkowej informacji: długie, parogodzinne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, bardzo dokładna analiza z Biurem Legislacyjnym, wiele pytań, wiele wątpliwości.

Dziękuję bardzo panu posłowi. I teraz przystąpimy do przedstawienia stanowisk klubów i koła. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Piotr Kaleta, który zaprezentuje stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo!

W ostatnich kilku latach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie orzekał na temat stosowania przepisów tejże dyrektywy. Dodatkowo projekt tej ustawy dostosowuje przepisy polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii Europejskiej. Ponadto projekt ustawy przewiduje wprowadzenie uregulowań pozwalających na zamieszczenie na kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu stosownych adnotacji oraz obrazu linii papilarnych.

Dlatego prosimy Wysoką Izbę także o poparcie tego projektu. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Dziękuję bardzo panu posłowi. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi pan poseł Michał Gramatyka. Wysoka Izbo! Tradycyjnie ustawa trafia pod obrady w ostatnim momencie i tradycyjnie Sejm nie dał posłankom i posłom czasu na dokładne zapoznanie się z jej projektem. Gdybyśmy chcieli li tylko przeczytać całość tego materiału, to nie starczyłoby nam na to 3,5 godziny, czyli tego czasu, w jakim obradowała wczoraj Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Nieco niejasne jest użycie klauzul generalnych, np.: można wydalić obywatela Unii z Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie względów obronności i bezpieczeństwa państwa. te klauzule generalne nie są zdefiniowane, a w naszej ocenie powinny być zdefiniowane. W zasadzie nie budzą też wątpliwości nowe uprawnienia dla funkcjonariuszy straży granicznych, chociaż sprawdzanie przez funkcjonariuszy, czy małżeństwo jest czy nie jest fikcyjne, przyznają państwo, ma aspekt nieco humorystyczny. Wysoka Izbo! Bardzo ciekawym wątkiem w procedowaniu nad tą ustawą jest jedna z przyczyn jej uchwalenia, czyli orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mój przedmówca poruszał zresztą ten wątek. Dwa z wielu przywołanych orzeczeń dotyczą Polaków: pani Szei i pana Ziółkowskiego. Przytaczam nazwiska dlatego, że w orzecznictwie TSUE nazwiskami oznacza się numery spraw, więc one i tak są publiczne. Oboje starali się o prawo pobytu w Niemczech, oboje dowodzili swojego prawa na podstawie nowatorskiej na tamte czasy przesłanki, która zakłada, że prawo stałego pobytu przysługuje każdemu obywatelowi Unii Europejskiej, który w danym kraju spędził legalnie 5 lat. W obu przypadkach lokalne sądy odmawiały Polakom uznania ich racji, podnosząc, że wskazane przez nich 5-letnie okresy rozpoczęły się w czasie, kiedy Polska nie była jeszcze członkiem Wspólnoty. W unijnej nowomowie oznacza to po prostu, że byli oni klientami niemieckiej opieki społecznej. Proszę sobie wyobrazić, że w obu tych przypadkach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał rację Polakom. W uzasadnieniu podnosił m.in., że nie można dzielić obywateli Unii Europejskiej na lepszych i gorszych tylko dlatego, że kraje nowej Unii uzyskały członkostwo później niż kraje starej Unii, że nie można rozróżniać obywateli Unii na tych bardziej albo mniej majętnych, że wszyscy w Unii jesteśmy równi. Tak właśnie działają wartości Wspólnoty Europejskiej, tak właśnie działa w Unii praworządność. Francuski sędzia w obronie polskich obywateli sprawozdawał wbrew stanowisku niemieckich sądów. Dla prawnika niektóre tezy tych uzasadnień są po prostu imponujące. Stopień uprawnień obywatela Unii nie wynika z czasu, jaki jego kraj jest członkiem Wspólnoty. Stopień tych uprawnień nie ma też nic wspólnego z sytuacją materialną tego obywatela. Dlaczego dzisiaj o tym mówię? Bo odnoszę wrażenie, że to są właśnie wartości, które państwo - kieruję te słowa do przedstawicieli rządu - kwestionują. Grozicie zawetowaniem unijnego budżetu, chcecie popchnąć Polskę na drogę prowadzącą do opuszczenia Wspólnoty. Przykładacie rękę do scenariusza dla naszej ojczyzny pisanego cyrylicą. To nie jest dyskusja o unijnym budżecie, o „Krajowym planie odbudowy i wzmocnienia odporności” To nie jest tylko kwestia miliardów, które możemy stracić, tu nawet nie chodzi o inne nasze uprawnienia, o wspólny rynek, o studentów, którzy pobierają edukację na europejskich uczelniach w ramach Erasmusa. To jest kwestia zasad, które leżą u podstaw funkcjonowania europejskiej Wspólnoty, to jest walka o idee, które są wypracowane przez Schumana, Adenauera, Spaaka czy Gasperiego. To jest walka o spuściznę naszych polityków: z Władysławem Bartoszewskim, Janem Kułakowskim czy panem prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Trawestując myśl ks. Jana Twardowskiego, którą przytoczył ostatnio pan prof. Michał Romanowski w jednym ze swoich felietonów: spieszmy się kochać Polskę w Unii Europejskiej. Tak krucha jest to wartość i tak szybko możemy ją stracić przez wasze nieodpowiedzialne działania. Dziękuję bardzo. W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy głos zabierze dwóch panów posłów: najpierw pan poseł Rafał Adamczyk, a następnie pan poseł Jan Szopiński. Panie Marszałku! Panowie Posłowie! Panie Dyrektorze! Panie Wiceministrze! Mieliśmy wczoraj niebywałą przyjemność kolejny raz procedować na hura nad kilkuset stronami projektu ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Proszę teraz pana posła Jana Szopińskiego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rada Ministrów uznała ten projekt za pilny z uwagi na konieczność uregulowania zasad wjazdu i pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin. Natomiast proszę o wyjaśnienie, dlaczego posłowie otrzymali 2 dni na przeczytanie tego dzieła, które ma bez mała 500 stron - to po pierwsze. Po drugie, czy regulacje brytyjskie zostały podane dopiero tak późno i w związku z tym jest nadane takie tempo pracy? Jaki jest powód tego, że po raz wtóry Wysoka Izba zostaje przymuszona do pracy nad dokumentem w tempie iście ekspresowym?

Aby poprawić jakość prowadzonych postępowań administracyjnych, wprowadziliście państwo do tej ustawy, która miała dotyczyć wjazdu i pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, jeszcze wiele innych uregulowań, tak jak zawsze, bo to się robi tak przy okazji. W związku z tym mam takie pytanie. Aby poprawić jakość prowadzonych postępowań administracyjnych, w projekcie ustawy wprowadza się przepis, który pozwala Straży Granicznej na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz sprawdzenie w miejscu pobytu obywatela Unii Europejskiej w przypadku podejrzenia zawarcia fikcyjnego małżeństwa. Dla Straży Granicznej wprowadza się określone regulacje, które określa się pod nazwą: prawdopodobieństwo. W związku z tym mam pytanie, na podstawie jakich przesłanek mogą powstać wątpliwości funkcjonariusza, czy małżeństwo jest fikcyjne, kto stwierdza taką wątpliwość i jak jest ona uzasadniona, jaką ma moc prawną.

Czy po wprowadzeniu zmian nie nastąpi dublowanie zadań Policji i Straży Granicznej w zakresie kontroli spraw pobytowych cudzoziemców na terenie Polski? Czy rozszerzenie kompetencji Straży Granicznej oznacza, że Policja dotychczas nie wywiązywała się z zadań, które dotyczyły weryfikacji małżeństw cudzoziemców? Kolejna kwestia. Mówiłem już o tym na posiedzeniu komisji. Mamy dualizm ustawowy, bo przypomnę Wysokiej Izbie, że Wysoka Izba przegłosowała na wniosek PiS-u takie regulacje, które umożliwią zatrudnianie w Polsce z jednej strony lekarzy, z drugiej strony pielęgniarek na podstawie dyplomu uzyskanego w krajach spoza Unii Europejskiej i oświadczenia na piśmie, że ten ktoś zna język polski. W związku z powyższym mam pytanie: Czy te regulacje, które zostały tak opisane, a przeciwko którym (Dzwonek) protestowały Naczelna Rada Lekarska i związek pielęgniarek i położnych, zostały zawarte również w regulacji z druku nr 798? Dziękuję. Dziękuję bardzo.

Dzień dobry, panie marszałku, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak jest. Panie Marszałku! Szanowni Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Koalicja Polska - PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści przedstawić stanowisko w odniesieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, który został zawarty w druku sejmowym nr 798. Szanowni Państwo! Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie tego projektu na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, można powiedzieć, w ekspresowym tempie. Ze względu na obszerność dokumentu nie dawało to możliwości wnikliwego przeanalizowania zawartych treści i proponowanych zmian. Zresztą wspominali już o tym moi przedmówcy. Projekt ustawy przybrał formę projektu pilnego z uwagi na konieczność uregulowania zasad wjazdu i pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin po okresie przejściowym wynikającym z ustawy o wystąpieniu ww. państwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, który kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.

Termin ten jest oczywiście nierozerwalnie związany z zakończeniem okresu przejściowego dla obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin.

Chciałam również powiedzieć, że z dniem 2 sierpnia 2021 r. wejdą w życie zasady wydawania zaświadczeń o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej, kart pobytowych, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu oraz kart stałego pobytu. Szanowni Państwo!

Sprawia to, że zostaną ujednolicone formaty dokumentów wydawanych obywatelom i że będą umieszczone adnotacje o stałym pobycie oraz obraz linii papilarnych. Z uwagi na krótki czas analizy i okres dostosowania do wejścia w życie projektu ustawy rodzi się wiele pytań w odniesieniu do kosztów wprowadzenia, wdrożenia w życie tej ustawy, a także nowych uprawnień Straży Granicznej w zakresie zaistnienia podejrzenia zawarcia fikcyjnego małżeństwa z obywatelem Unii Europejskiej, o czym również przed chwileczką wspominał mój przedmówca. Straż Graniczna na podstawie nowych uprawnień ma przeprowadzać wywiad środowiskowy oraz dokonywać sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela Unii Europejskiej, czy nie zaistniało podejrzenie i czy to podejrzenie jest uzasadnione.

Decyzja o wydaleniu tych obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin będzie wydawana, z urzędu bądź na wniosek, przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, a nie - jak do tej pory - przez wojewodę. Szanowni Państwo! Reasumując (Dzwonek), potrzeba wprowadzenia tej ustawy jest zrozumiała, ale w trosce o pracę funkcjonariuszy Straży Granicznej i wykonywane rzetelnie przez nich obowiązki chciałam zapytać, czy rzeczywiście wdrożenie w życie tej ustawy jest na tyle mocno zaawansowane, że ci funkcjonariusze będą mieli wszystkie instrumenty do sprawnego prowadzenia zlecanych zadań, i czy rzeczywiście wszystkie te mechanizmy, środki i koszty będą im zapewnione. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę teraz pana posła Krzysztofa Tuduja, który w imieniu koła Konfederacja przedstawi stanowisko. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozmawiamy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, wprowadzenia instytucji cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej oraz uregulowania nowych podstaw prawnych dotyczących odmowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu, a także stosowania przez Polskę umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej w przypadku praw pobytowych obywateli brytyjskich i członków ich rodzin. Sama nazwa i zakreślenie przedmiotu ustawy są bardzo rozbudowane, podobnie jak sam projekt, który wraz z uzasadnieniami liczy prawie 700 stron, o czym tutaj już było wspomniane. Omawiana regulacja ma charakter dostosowania polskich przepisów w następujących obszarach: przemieszczania się i pobytu w Unii Europejskiej, rozwiązań dotyczących uprawnień Straży Granicznej. Dostosowanie ma miejsce również w obszarze umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Większość tych rozwiązań ma wejść w życie już 1 stycznia 2021 r., stąd pośpiech w procedowaniu nad tą ustawą. Przy tej okazji chciałbym wspomnieć wyznawcom wiary stanowiącej, że nie ma zbawienia poza Unią Europejską, że ta regulacja w kontekście Wielkiej Brytanii powinna przypomnieć, że można kształtować swoje stosunki międzynarodowe nie tylko grupowo, ale również bilateralnie. Wielka Brytania prowadzi własną politykę w oparciu o swoją ocenę korzyści i kosztów w relacjach międzynarodowych, w oparciu o jak najlepsze pojęcie własnego interesu. Tak powinno postępować każde szanujące się państwo. Można i koniecznie trzeba walczyć o polskie interesy, będąc wewnątrz Unii Europejskiej, ale jak pokazuje przykład brytyjski, można realizować własną politykę również w inny sposób. My jako państwo polskie powinniśmy mieć przemyślane i przygotowane różne strategiczne scenariusze, różne warianty postępowania, bez eliminowania opcji przygotowania bezpiecznego wyjścia awaryjnego, właśnie ze względu na bezpieczeństwo, na wypadek, gdyby wystąpiło ryzyko, że w Unii Europejskiej będziemy się dusić, gdy taki klimat polityczny i prawny stworzą nam lewicowe kręgi zarządzające Unią Europejską. Przyszłość może wyglądać różnie, trzeba być gotowym na każdy wariant. Wreszcie taki scenariusz powinien być przygotowany również jako argument negocjacyjny w różnych toczących się dyskusjach w ramach pilnowania polskich spraw, kiedy się jest w Unii Europejskiej. No, do tego potrzebna jest wyobraźnia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa posłów chciałby jeszcze dopisać się do listy osób chętnych do zadania pytania? Jeżeli nie, to zamykam tę listę, ustalając czas na zadanie pytania - 1 minuta. Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W projekcie ustawy jest dużo ogólnych sformułowań, które mogą prowadzić do daleko idącej swobody w podejmowaniu decyzji. Jako przykład podam stwierdzenie: obywatel Unii Europejskiej posiada wystarczające środki finansowe. Brak doprecyzowania, co to oznacza. Kolejne: według jakich kryteriów należy badać, czy życie rodzinne z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej zostało rozwinięte lub umocnione? Tutaj również decyzje będą podejmowane indywidualnie. Moja obawa jest taka: Czy nie będzie problemu z zastosowaniem tej ustawy? Czy nie nastąpi zablokowanie urzędów wojewódzkich, tak jak jest obecnie, przy rozpatrywaniu spraw cudzoziemców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej? To, co się dzieje w urzędach [[Dzwonek]] wojewódzkich, to jest po prostu tragedia, tak długo oczekuje się na rozpatrzenie sprawy. Dziękuję bardzo. Pytanie teraz zada pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Procedowany projekt jest oczywiście bardzo obszerny, zawiera regulacje odnoszące się m.in. do uprawnień Straży Granicznej czy do stosowania umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii, ale nie zawiera jednej, wydaje mi się, istotnej - a może dla rządu nieistotnej - regulacji. To jest regulacja, w sprawie której się zwracałem już do ministerstwa spraw wewnętrznych, a mianowicie regulacja dotycząca nieformalnych związków partnerskich par dwunarodowościowych. Problem polega na tym, że jeżeli taka para nie zawarła związku małżeńskiego, to obecne regulacje pandemiczne nie pozwalają tym osobom na kontynuowanie wspólnego pożycia ze względu na to, że są obywatelami innych krajów, oczywiście w przypadku gdy jedna z osób jest obywatelem spoza Unii Europejskiej. Przepisy umożliwiające taki wspólny pobyt już wprowadziły m.in. Czechy, Dania, Norwegia, Holandia, Austria czy Szwajcaria. W tym miejscu też warto zaznaczyć, że Polacy zdecydowanie są za Unią i mówią: tak dla Unii, nie dla weta. Natomiast pamiętajcie, że miłość to nie turystyka.

Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zadanie pytania panią poseł Joannę Fabisiak, Koalicja Obywatelska.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dwa pytania. W sprawozdaniach i wypowiedziach słyszałam głównie o relacjach z Wielką Brytanią, co jest naturalne, bo od stycznia ta sytuacja się zmieni. Ja chciałabym spytać o inny kierunek, a mianowicie o Ukrainę. Bardzo wielu obywateli polskich, którzy nabyli obywatelstwo w drodze Karty Polaka, przyjeżdża do Polski. Myślę tu głównie o kobietach, które są bardzo potrzebne, to są panie, które są często ze starszymi osobami, opiekują się starszymi osobami.

Chciałabym prosić o odpowiedź i o odpowiedź na piśmie. Wydaje mi się, że te regulacje mogą bardzo utrudnić relacje wzajemne w sumie Polaków czy też Polek, które tu pracują, z ich współmałżonkami i rodzinami. Z tego, co wiem (Dzwonek), te rodziny bardzo często przyjeżdżają i chcą przyjeżdżać, i chcą, żeby te relacje były wzajemne. Tymczasem to Straż Graniczna teraz będzie oceniała, czy to jest małżeństwo, czy mogą przyjechać itd. Nie otrzymałam. To bardzo duża ustawa, nowelizacja ustawy, implementacja prawa europejskiego, ale nie ma zarządzenia. A jakie jest to zarządzenie? Czy ono jest gotowe? Dziękuję, pani poseł. Nie widzę na sali pana posła Mirosława Suchonia. Zatem proszę o zadanie pytania pana posła Wojciecha Saługę. Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Sejm ma podejmować prace i pracować nad ustawami, a jesteśmy przymuszeni do tego, żeby 500 stron procedować w 2 dni. Tego nie da się ani przeczytać, ani zrozumieć, a już nie mówię, jakieś poprawki wnieść. A na koniec - to się tyczy tysięcy naszych obywateli i członków ich rodzin. To jest życie ludzi. I tak gramy życiem ludzi, że uchwalamy na kolanie przepisy w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie ich przeczytać. Chciałem zapytać o te klauzule generalne, o wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względów obronności, bezpieczeństwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego. To wszystko fajnie brzmi. Chciałem spytać, kto o tym będzie decydował, ponieważ będą to rzeczy bardzo uznaniowe, a jak są uznaniowe, to jest absolutna dowolność. Czy nie ma szans tego po prostu [[Dzwonek]] zawęzić, nazwać, skatalogować, żeby ludzie wiedzieli, na czym stoją i czego się mogą trzymać? Dziękuję bardzo. Pytanie zada teraz pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Przewodniczący Komitetu Kaczyński! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Debatujemy o swobodnym przemieszczaniu się w Unii, jednak już niedługo może nas to nie dotyczyć. A ja chciałabym wyrazić wdzięczność parlamentowi holenderskiemu za to, że zajął się kwestią łamania praworządności w Polsce. Przypomnę, że wezwał on swój rząd do postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niewykonywanie wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Od 5 lat ta izba daje przyzwolenie na dewastację prawa, najpierw w Polsce, a teraz już w całej Unii Europejskiej. Marszałek Witek, tu nie ma się co dziwić. Tu trzeba przepraszać za to, że w obliczu takiego nieszczęścia Polska teraz blokuje pomoc dla chorych i cierpiących sióstr i braci w całej Unii Europejskiej. Co to za szatański pomysł, żeby w ten sposób karać bezbronne narody? Wy nie macie ludzkich uczuć. Nie wiecie, co to empatia i współczucie. Wstydzę się dzisiaj za ten Sejm, wstydzę się za ten rząd i dzisiaj przez was wstydzę się, że jestem Polką. Dziękuję bardzo.

Wielka Brytania wprowadziła system punktowy dla obywateli Polski i innych krajów Unii Europejskiej, którzy zamierzają przebywać w niej dłużej niż 6 miesięcy. Czyli de facto Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będzie blokowało na swoim terenie pobyt dużej grupy Polaków i realizowało typowy drenaż mózgów i specjalistycznych kadr. Mam pytanie do przedstawicieli rządu: Czy polski rząd rozważał wprowadzenie na zasadzie wzajemności takich samych zasad uzyskiwania prawa pobytu obywateli Wielkiej Brytanii na terenie Polski, jakie rząd Wielkiej Brytanii wprowadził wobec obywateli Polski? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Korzystając z okazji swobodnego przemieszczania się członków obywateli Unii Europejskiej, chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć to, co dzieje się w Polsce. Otóż państwo zamknęliście praktycznie całą branżę turystyczną. Dzisiaj na południu Polski od Karkonoszy po Zakopane 80% podmiotów, głównie rodzinnych, prywatnych, polskich jest zamkniętych przez to, że od 14 października nie pozwalacie ludziom na normalne funkcjonowanie. Jeżeli zamykacie branżę, nie dajecie żadnych rekompensat. Dlatego apelujemy, po pierwsze, o to, aby znalazła się pomoc dla branży turystycznej, dla branży gastronomicznej, dla tych wszystkich ludzi, którzy przez lata inwestują, abyśmy mogli w normalny sposób spędzić okres ferii. Niezbędne jest to, aby wydłużyć także ten sezon ferii (Dzwonek), aby pozwolić na bezpieczne ich spędzenie, a tysiącom Polek i Polaków pozwolić na to, aby przetrwali w COVID-zie do czasu sezonu letniego. Dziękuję bardzo panu posłowi. Na zadane wcześniej pytania odpowiedzi udzieli szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców pan Jarosław Szajner.

Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Jak już panowie, panie posłanki, jak państwo wskazywaliście, ta ustawa jest niezbędna do przyjęcia, abyśmy mogli w sposób jak najbardziej prawidłowy zapewnić możliwość życia i funkcjonowania u nas obywateli Wielkiej Brytanii, jak również poprawić bezpieczeństwo dokumentów posiadanych przez obywateli Unii Europejskiej. Chciałbym krótko odpowiedzieć na pytania. Może zacznę od pytań pana posła Szopińskiego. Tak, rozważaliśmy wiele wariantów. Został wybrany wariant najlepszy, wariant, który jest jak najbardziej odpowiedni ze względu na liczbę obywateli Wielkiej Brytanii przebywających w Polsce, jak też jak najbardziej korzystny dla naszego kraju.

Jeżeli chodzi o sytuację odnośnie do wywiadu środowiskowego. To dotyczy tego, czy Straż Graniczna jest przygotowana - pani poseł Nowogórska zadała to pytanie - do przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Tak, jest przygotowana. Takie wywiady też przeprowadzają w sytuacji, które dotyczą obywateli państw trzecich. Jeżeli chodzi o sytuację lekarzy i pielęgniarek, to akurat ta sytuacja w ogóle nie ma związku z tą ustawą, ponieważ oni nabywają prawo pobytu w związku z podejmowaniem pracy, a nie w związku z zawieraniem małżeństwa.

Koszty są podane w ocenie skutków regulacji. Jest to koszt dostosowania systemów i koszt blankietów do wydawania kart.

Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Saługi odnośnie do sformułowań generalnych, ogólnych i o to, kto podejmuje decyzje o wydaleniu obywatela Unii Europejskiej, to jest to jasne. Trzeba też wziąć pod uwagę, że od tej decyzji jest możliwość odwołania do sądów administracyjnych. Na pozostałe pytania odpowiem na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Nie ma. Zatem zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw (druki nr 799 i 820) Bardzo proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Ministrze! Komisja Finansów Publicznych na wczorajszym posiedzeniu rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw, druk nr 799. Odbyło się pierwsze czytanie tej ustawy. Pierwsza wersja specustawy funduszowej wprowadziła regulacje, których celem była płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych w warunkach kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19.

Podczas posiedzenia komisji omówiono szczegółowo poszczególne zmiany zawarte w projekcie ustawy i zgłoszono dwie poprawki. Komisja Finansów Publicznych w głosowaniu obie poprawki zaopiniowała negatywnie. W imieniu Komisji Finansów Publicznych wnoszę do Wysokiej Izby o uchwalenie rzeczonego projektu ustawy, a na żądanie wnioskodawców poprawki komisja przedstawia wniosek mniejszości polegający na skreśleniu w art. 1 pkt 3. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Przystępujemy teraz do przedstawienia stanowisk klubów i koła. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Teresa Pamuła, która zaprezentuje stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość stanowiska dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw, druk nr 799. Szanowni Państwo! Tak jak już wspomniał poseł sprawozdawca, projektowana ustawa wprowadza nowe regulacje mające usprawnić działania zmierzające do przezwyciężenia konsekwencji gospodarczych i społecznych spowodowanych stanem pandemii. Specustawa funduszowa wprowadza regulacje, których celem byłaby płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych w warunkach kryzysu wywołanego pandemią.

Projekt ustawy pozwala na rozszerzenie też w zakresie funduszy ustawy funduszowej z zastosowaniem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Włączenie tych programów w ramach tego instrumentu da podstawę prawną do tego, aby skutki COVID-owskie miały mniejsze oddziaływanie na ustawę. Projekt ustawy zakłada także nowelizację ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, wprowadzając do przepisów sprawy z zakresu opracowania planów rozwojowych. Z kolei nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju umożliwia realizację polityki Unii Europejskiej w zakresie łagodzenia społecznych i gospodarczych skutków kryzysu wywołanego przez pandemię. Projekt przewiduje wzmocnienie kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako odpowiedzialnego za przygotowanie planu rozwojowego stanowiącego podstawę do ubiegania się o środki uruchamiane w celu łagodzenia skutków kryzysu i uniknięcia pogłębiania się nierówności w Unii Europejskiej. Bardzo istotne jest, aby regulacje zapewniały w ramach planu rozwoju wsparcie stanowiące pomoc publiczną zgodną z przepisami unijnego prawa materialnego i proceduralnego w tej dziedzinie. Projekt przewiduje także nieuwzględnianie przy wyliczaniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej wydatków i kosztów, które zostały pokryte ze środków finansowych pochodzących z programów finansowanych lub dofinansowanych ze środków funduszy europejskich, programów krajowych czy też dotacji z budżetu państwa.

Projektowane przepisy umożliwią ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego przygotowanie programu finansowanego właśnie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt ustawy, co jest bardzo istotne, nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, jak również będzie oddziaływał pozytywnie na rynek pracy, i zwiększa stabilizację wśród przedsiębiorców i da możliwość zatrudniania na dotychczasowym poziomie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw jest bardzo ważny, ponieważ czekają na niego beneficjenci programów realizujących projekty ze środków unijnych, pracodawcy, pracownicy, instytucje uczestniczące w systemach wdrażania środków europejskich, podmioty prowadzące domy społeczne, a takich podmiotów jest przeszło 800, osoby ponoszące płatność za społeczne domy pomocy, czyli prawie 80 tys. osób. Dziękuję bardzo. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi pani poseł Paulina Hennig-Kloska. Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej w sprawie ustawy wspierającej realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., która jest przedłużeniem ustawy przyjętej przez nas na wiosnę tego roku i wprowadza poluzowanie zasad wydatkowania i rozliczania środków europejskich w Polsce. Tak się składa, że ta nowelizacja dotyczy środków europejskich zarówno w obecnej, jak i w przyszłej perspektywie. Jest to dokument rządowy, pod którym podpisał się, jak rozumiem, również pan premier Mateusz Morawiecki.

I chciałam przy tej okazji zapytać: Które stanowisko rządu premiera Morawieckiego jest prawdziwe? Czy to, że środki europejskie nie są nam potrzebne, a tym bardziej - pilnie potrzebne, że możemy sobie bez nich poradzić, wyjdziemy z kryzysu cało, a w ogóle to mamy takie same w tej samej cenie albo i tańsze środki dostępne w ramach własnych możliwości, czy to, że jednak te środki europejskie są potrzebne, by walczyć z ubożeniem społeczeństwa, które może być następstwem właśnie obecnego kryzysu epidemiologicznego, który przeżywa cały świat?

No nie, prawda jest taka, że Polska wciąż nie jest płatnikiem netto w Unii Europejskiej i wyciąga z tej Unii więcej w ramach corocznych zaliczek niż wpłaca do kasy unijnej, bo wciąż należymy do krajów rozwijających się, goniących średnią PKB w Unii Europejskiej. W związku z czym środki, które mogą być dla nas przeznaczone, to jest 750 mld w ramach funduszu odbudowy, na które czekają polscy przedsiębiorcy i obywatele, i z części budżetowej Unii Europejskiej. Są nam one pilnie potrzebne i będą dużym dodatkiem do tych możliwości, z których Polska na co dzień korzysta.

Szacuje się m.in., że te, które będą wyemitowane, będą mniej więcej 2 punkty procentowe tańsze od tego, co możemy my uzyskać.

Niech mi pan uwierzy, Unia Europejska ma dużo tańszy dostępny pieniądz i nie ma potrzeby, żebyśmy corocznie jeszcze więcej miliardów płacili z powodu odsetek, płacili z naszych kieszeni, kieszeni podatników, bo wam się tak podoba, bo macie konflikty wewnętrzne, bo Morawiecki walczy z Ziobrą, bo politykę własnej partii i własnego rządu przedkładacie nad interes narodowy, interes obywateli i polskiej gospodarki. Nie ma na to naszej zgody i nigdy nie będzie.

Ustawa oczywiście, jak powiedziałam, luzuje wydatkowanie środków europejskich, co z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne i istotne, jak również rozliczanie tych środków oraz wprowadza nowe fundusze. Będziemy ją oczywiście popierać. Bardzo dziękuję, pani poseł. W imieniu klubu Lewica głos zabierze pani poseł Anita Sowińska. Zatem w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści głos zabierze pan poseł Krzysztof Paszyk. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Chciałbym na wstępie zadeklarować, że oczywiście Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści będzie popierał ten projekt, bo na sercu leży nam to, aby wszelkie procedury związane z rozliczaniem funduszy europejskich, z ich docelowym dotarciem bez przeszkód się zrealizowały.

Po pierwsze, wiosną ubiegłego roku procedowaliśmy nad podobnymi rozwiązaniami.

Z uporem maniaka, absolutnie, na zasadzie wyłączności waszej wiedzy, dogmatu waszej doskonałości i wiedzy nie chcieliście o tych rozwiązaniach słuchać. To jest pierwsza rzecz, za którą ja bym się na pańskim miejscu nieco wstydził.

Środki europejskie są niezwykle potrzebne nie tylko polskim samorządom, polskim przedsiębiorcom, polskim rolnikom, ale też naszej gospodarce. Środki z funduszu odbudowy są niezbędne, potrzebne, abyśmy ustabilizowali niezwykle rozchwianą dzisiaj służbę zdrowia, zorganizowali ją na nowo. Tego się bez funduszy europejskich zrobić nie da i warto wykorzystać tę okazję, tę debatę, którą dzisiaj prowadzimy, aby to jasno wybrzmiało.

Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę teraz pana posła Michała Urbaniaka, który przedstawi stanowisko Koła Poselskiego

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W porządku, ja to wydłużenie zasadniczo rozumiem, to jest usprawiedliwione, ponieważ kryzys, który teraz mamy, jest kryzysem, który w wielu aspektach trudno przewidzieć. Natomiast czy wy jako rządzący, państwo z rządu tzw. dobrej zmiany, zamierzacie dalej trzymać Polaków niemal pod ścianą w sprawach gospodarczych, w sprawach edukacji czy w sprawach kulturalnych?

Piloci wycieczek czy przewoźnicy, którzy też przez was nie mogą pracować, za chwilę wywiozą was na taczkach. I co, dalej będziecie mówić, że ratujecie gospodarkę? Czy premier Morawiecki dalej będzie mówić o tym, że dla niego każde miejsce pracy jest na wagę złota? Po czym zamyka stocznię Gryfia. Polacy nie są tak naiwni, jak się wam wydaje, i Polska już długo tak nie pociągnie. Na dodatek chcecie sobie po prostu na Polakach poeksperymentować. Jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, by w Polsce była wysoka zaszczepialność na różne choroby, natomiast w momencie gdy mamy produkty, które jeszcze nie są dostatecznie dobrze przebadane, które jeszcze powinny być testowane, wy w praktyce - bo w teorii tak nie będzie, ale w praktyce tak będzie - będziecie próbować wymusić na Polakach to, aby przyjmowali takie substancje. Kto weźmie za to odpowiedzialność? Bo myślę, że wy umyjecie ręce. Poza tym, biorąc pod uwagę wydolność naszego systemu ochrony zdrowia, zaszczepienie choćby połowy populacji w Polsce może zająć ponad 3 lata. Może minister Niedzielski jest magikiem, może jest w stanie zrobić to jakoś szybciej, ale czary raczej nie istnieją. Jeśli ma się to wiązać z dalszym tresowaniem Polaków, to zwiększaniem, to zmniejszaniem po prostu obostrzeń, stwierdzaniem na podstawie sondaży, że teraz lepiej trochę przycisnąć śrubę, a potem trochę ją odpuścić, to państwo od dobrej zmiany w przyszłym parlamencie już się nie znajdziecie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Czy pojawiła się może pani poseł z Lewicy, aby zaprezentować stanowisko? Nie. A zatem informuję, że lista posłów zapisanych do zadania pytania została zamknięta. Czas na zadanie pytania wyznaczam na 1 minutę. Proszę bardzo. Wysoki Sejmie! Chciałam zapytać, jakie jest zagrożenie, jeśli chodzi o niewykorzystane środki unijne z obecnej perspektywy finansowej, gdy rozporządzenie w sprawie tzw. praworządności wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku. Czy te środki, które są tak bardzo potrzebne polskiej gospodarce, przedsiębiorcom, samorządom, nie zostaną zablokowane? Polacy bardzo potrzebują funduszy unijnych. Tak dla Unii, nie dla weta. Dziękuję bardzo. Pytanie zada teraz pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej Polska zyskała gigantyczne środki finansowe wspomagające rozwój kraju, które przyczyniły się do niwelowania różnic w poziomie życia w Polsce i w krajach zachodniej Europy. W tym projekcie ustawy luzujecie formułę finansową dla wykorzystania tych środków - i bardzo dobrze - twierdząc, że przyczynią się one do szybszego usunięcia skutków kryzysu wywołanego COVID-19. To jak to jest w końcu: środki europejskie pomagają, czy nie pomagają? Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To, że od marca walczymy z koronawirusem, jest dla wszystkich oczywiste. I oczywiste również dla wszystkich było to, że będą problemy, że nie uda się rozliczyć części tych projektów dofinansowanych z programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Największym problemem jest to, że powołujecie się na unijną perspektywę, nową unijną perspektywę budżetową. W związku z tym przede wszystkim należy zapytać: Czy zdecydowaliście się finalnie zawetować budżet europejski i pozbawić Polskę miliardów złotych? Czy w przypadku szaleńczego weta prowizorium budżetowe pozwoli zrealizować założenia projektowe? Dziękuję serdecznie. Pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska, klub parlamentarny. Jest pan poseł Suchoń? Pan poseł Krzysztof Gadowski. Dobrze, że jest pan poseł Krzysztof Gadowski, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Robicie to teraz. Jaka jest przyczyna wprowadzenia tych programów w ramach tego instrumentu sąsiedztwa? Oczywiście ta ustawa przedłuża swoją działalność do tego, co oczywiście jest i będzie wchodziło. Pytanie następne: Czy państwo przewidujecie wprowadzenie podobnych mechanizmów do użycia w przypadku uchwalenia Funduszu Odbudowy i przyjęcia projektu budżetu Unii Europejskiej? Czy będzie można również tamte środki finansowe sprawnie wykorzystać i sprawnie poprowadzić inwestycje w ramach środków, które otrzymamy?

Dziękuję. Pan poseł Tomasz Piotr Nowak, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Jeżeli się nic nie zmieniło. Witam serdecznie pana marszałka, witam pana ministra, panów. Wysoka Izbo! I to powtarzali z pełnym przekonaniem posłowie PiS-u. W związku z tym proszę mi powiedzieć, czy jeśliby było wprowadzone prowizorium budżetowe, toby zlikwidowano takie programy, jak „Horyzont Europa”, „Unia Europejska dla zdrowia”, Europejski Fundusz Obronny, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, fundusz zarządzania granicami, Erasmus, „Kreatywna Europa”, LIFE+ itd., itd. Nie można posuwać się w swoich narracjach tak daleko, że po prostu ludzi traktuje się jak ciemną masę. Jest granica propagandy. Wydaje się, że wszyscy - badania to pokazują - jesteśmy euroentuzjastami, ale racjonalnymi euroentuzjastami (Dzwonek) i wiemy doskonale, że jutro trzeba powiedzieć: tak dla Unii Europejskiej, nie dla weta. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Joanna Fabisiak.

Proszę bardzo, pani poseł. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pierwsze pytanie. Mamy prolongować ustawę, która za miesiąc wygasa, więc mam pytanie. Tymczasem mówimy teraz, że są szczepienia, że prawdopodobnie sytuacja się poprawi już latem. Takie są przewidywania.

Im więcej specustaw, tym mniejsza rola parlamentu. To nie jest dobre i to powinno być inaczej rozwiązywane nawet w obecnej sytuacji, która nie jest do końca przewidywalna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Dariusz Klimczak, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Tak działo się w każdym regionie, także w moim. Chciałem zapytać o inicjatywę dotyczącą budowy 100 obwodnic. Czy państwo. Nie dostałem niestety jeszcze odpowiedzi na moją interpelację, a państwo dzisiaj tutaj są.

W jaki sposób chcecie państwo kontynuować budowę 100 obwodnic? Dziękuję bardzo.

Panie i Panowie Posłowie! Przede wszystkim: tak dla Unii, nie dla weta.

Przewiduje się, że społeczeństwo będzie na skutek kryzysu niestety ubożeć i musimy temu przeciwdziałać. Czy prawdą jest, panie ministrze, że weto przed niczym nas nie chroni, skoro nie chcecie praworządności, a ona i tak przy prowizorium będzie obowiązywać. To niestety jest fakt.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Szlachta, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

Wysoka Izbo! Podczas emocjonalnej dyskusji nad tym ważnym projektem ustawy część posłów dokonała inwersji podmiotowej, jeżeli chodzi o projekt ustawy.

Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pana ministra Waldemara Budę o udzielenie odpowiedzi. Tak? To przy okazji odpowie sobie pan na to pytanie, które pan zadał. To będzie miłe. Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

można powiedzieć, że dokończenia obecnej perspektywy.

Natomiast te wszystkie rozwiązania techniczne, które dotyczą wydatkowania środków europejskich w związku z COVID-19 i uproszczenie wydatkowania tych środków dotyczą dokończenia tej perspektywy.

Dlaczego - bo tutaj takie zarzuty padały - w pierwotnej wersji ustawy w kwietniu była propozycja, żeby ta ustawa obowiązywała tylko do końca roku? Szanowni Państwo! Pamiętam takie głosy, z których wynikało, że państwo by mieli wątpliwości, dlaczego też tak długo.

Tu powinna być pełna zgoda w tym zakresie. Być może pokrótce należałoby się do tego odnieść, bo państwo nie rozumieją, że można z jednej strony lubić środki europejskie, a z drugiej strony twardo je negocjować. Godzenie się na dzisiejszą propozycję ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady jest godzeniem się na to, że te środki są po prostu zagrożone, byłyby zagrożone w kolejnej perspektywie.

W rankingach, jeśli chodzi o absorbcję środków europejskich, jesteśmy w czołówce.

Uznajmy, bo to jest bezsprzeczne, że 750 mld wynegocjowane przez pana premiera to rzeczywiście jest gigantyczna suma, to jest gigantyczny sukces z lipcowego posiedzenia Rady Europejskiej. Jednak nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze i utrata pewnej niezależności, suwerenności i swobody w podejmowaniu decyzji w wielu segmentach, które dzisiaj nie są objęte traktatami, nie jest warta tych środków i nie zawsze nawet w życiu prywatnym, w zwykłym życiu jesteśmy w stanie wszystko przeliczyć na pieniądze (Dzwonek) i powiedzieć, że zawsze one wygrywają. W związku z tym, szanowni państwo, bardzo dziękuję za debatę nad tą ustawą. Mam nadzieję, że parlament ją przyjmie, a co do poprawek, to oczywiście moja opinia wyrażona w komisji będzie taka, że to są poprawki, które nie zasługują na poparcie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Szlachta, sprawozdawca. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałem bardzo krótko mimo wszystko podziękować wszystkim klubom.

A więc ta warstwa może bardzo głośnych wystąpień pozamerytorycznych nie przykryła jednak celu podstawowego, aby polski parlament przyjął ten ważny projekt ustawy. Dziękuję panu. Może ustawa po prostu była dobra? Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

Żeby nie było, że tylko posłowie w tym budynku pracują. Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Marcina Warchoła o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Proszę bardzo, panie ministrze. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Celem projektu jest wdrożenie dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie praw pokrzywdzonych, w szczególności dzieci, przestępstwami wykorzystania seksualnego. Większość tych uprawnień mamy już dzisiaj w naszym Kodeksie postępowania karnego, natomiast doprecyzowujemy jedynie komplet tych uprawnień, jeśli chodzi o należytą informację dla takiego pokrzywdzonego. Ale o tym w drugim punkcie. Mamy kilkadziesiąt spraw rocznie z zakresu handlu ludźmi i często pokrzywdzeni, osoby małoletnie, trafiają bez dokumentów do naszego kraju jako ofiary handlu ludźmi lub innych przestępstw transgranicznych. Bardzo trudno jest ustalić ich wiek: nie mają żadnych dokumentów, nie ma żadnych dowodów, ile mają de facto lat. W tym momencie wprowadzamy domniemanie małoletności. Jeżeli organ procesowy bądź inny funkcjonariusz - Służby Granicznej czy Służby Celnej - nie będzie w stanie określić wieku takiego małoletniego pokrzywdzonego, przepis im pomoże. Jest domniemanie, że ten, kto wygląda jak małoletni, rzeczywiście jest małoletnim i korzysta z wszystkich uprawnień małoletniego pokrzywdzonego w danym postępowaniu karnym. Tak że to bardzo ważny pierwszy przepis.

Natomiast przepis, który wprowadzamy, zakłada wejście w dialog przez organ procesowy, czy to prokuratora, czy sędziego, z pokrzywdzonym i odebranie od niego informacji, czy rzeczywiście zapoznał się z tymi uprawnieniami, czy wie, co może w tym postępowaniu, czy rozumie udzieloną mu informację i wreszcie czy chce z tego skorzystać.

Organ odbierze od pokrzywdzonego oświadczenia, czy chce on zastosowania wskazanych tam środków ochrony i wsparcia pokrzywdzonego. Jakie to są środki? Chodzi tu m.in. o przesłuchanie pokrzywdzonego tylko raz. Bardzo często zdarza się, że małoletni pokrzywdzony czy pokrzywdzony pełnoletni nie jest w stanie w sposób należyty rozróżnić tego, jakie posiada uprawnienia.

Przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego, kuratora na odległość, utrwalenie czynności za pomocą obrazu i dźwięku, utajnienie danych świadka, wyproszenie z sali przesłuchań oskarżonego, żeby jego obecność nie wpływała krępująco na świadka, wyłączenie jawności postępowania, przesłuchanie świadka i oskarżonego na odległość - szereg tego typu uprawnień zwanych środkami ochrony będzie zagwarantowanych pokrzywdzonemu w sposób realny, a nie tylko poprzez wręczenie kartki papieru. Bardzo proszę Wysoką Izbę o poparcie tego projektu. Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubu i koła. Jako pierwszą zapraszam panią poseł Annę Milczanowską z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pragnę zaprezentować stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, druk nr 732. Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w Kodeksie postępowania karnego zmierzających do uściślenia i doprecyzowania przepisów regulujących uprawnienia procesowe pokrzywdzonych. Proponowana zmiana ma na celu uwzględnienie w wniosków Komisji Europejskiej dotyczących niepełnego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępujących decyzję ramową Rady, a także dyrektywy Parlamentu i Rady z grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej zastępującej decyzję ramową Rady z 2004 r. Rozważana treść art. 49b Kodeksu postępowania karnego ma za zadanie określenie wprost zasad postępowania w sytuacji, gdy istnieją wątpliwości co do wieku pokrzywdzonego w warunkach, w których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że jest on małoletni. Zgodnie z powyższą zmianą przepisów we wskazanych okolicznościach będą miały zastosowanie przepisy dotyczące małoletnich i pokrzywdzonych. Druga z proponowanych zmian nakłada na organ prowadzący postępowanie karne obowiązek zbadania okoliczności sprawy celem ustalenia właściwości warunków osobistych pokrzywdzonego. Powyższe ma służyć ochronie gwarancji procesowych pokrzywdzonego. Organ prowadzący postępowanie co do zasady będzie zobligowany zwrócić się do pokrzywdzonego celem odebrania od niego oświadczenia co do chęci skorzystania ze wskazanych w proponowanym przepisie instytucji mających na celu poprawę sytuacji pokrzywdzonego. Przepis ten ma na celu zaakcentowanie obowiązku indywidualnego podejścia do ofiary przemocy przez organ prowadzący postępowanie karne. Z uwagi na to, że proponowane zapisy mają na celu poprawę położenia pokrzywdzonych w toku postępowania karnego, a przyjęcie przepisów w przedstawionym kształcie ma służyć pełnemu i jednoznacznemu wdrożeniu dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za przyjęciem projektowanej ustawy w proponowanym brzmieniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Arkadiusz Myrcha, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie pośle, zapraszam pana serdecznie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy zmieniającej Kodeks postępowania karnego, zawartego w druku nr 732.

Sprawą oczywistą jest, że przedmiotem elementarnej odpowiedzialności każdego państwa jest zapewnienie czytelnych dla każdego uczestnika postępowania - czy to przygotowawczego, czy następnie sądowego - jasnych reguł postępowania, zwłaszcza w okolicznościach tak wrażliwych, jakie występują w przypadku popełnienia czynów zabronionych, gdzie osobą pokrzywdzoną jest osoba małoletnia. I istnieje pewna luka w przepisach Kodeksu postępowania karnego, nie określa się w sposób czytelny, jak organ powinien postępować w takich przypadkach. Przygotowana w związku z tym propozycja zmian w Kodeksie postępowania karnego wydaje się propozycją dobrą i zasługującą na poparcie. Dlatego Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska wnioskuje o przekazanie tego projektu do dalszych prac w komisjach. Będziemy oczywiście aktywnie w nich uczestniczyć.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Ueberhan, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu klubu Lewicy przedstawić stanowisko klubu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Jak czytamy w przedłożeniu, projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Przedłożony projekt wprowadza do Kodeksu postępowania karnego zmiany, które uściślają i doprecyzowują obowiązujące już obecnie przepisy odnoszące się do gwarancji procesowych przysługujących osobom pokrzywdzonym. Konieczność wprowadzenia tych zmian wiąże się z wykonaniem zobowiązań wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej.

W polskim prawie przepisy obecnie zawarte w Kodeksie postępowania karnego realizują już w większości postanowienia wskazanych wcześniej dyrektyw. Są to m.in. przepisy dotyczące prawa pokrzywdzonego do informacji o przysługujących mu uprawnieniach i do informacji na temat postępowania, prawa do tłumaczenia, w tym do złożenia zawiadomienia o przestępstwie w języku, którym włada pokrzywdzony, prawa do bycia wysłuchanym, do pomocy prawnej, do zwrotu poniesionych wydatków, do odszkodowania, do środków ochrony, a ponadto w Kodeksie karnym wykonawczym w zakresie dotyczącym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, mającym zapewnić środki pomocy dla pokrzywdzonych, w tym pomocy materialnej oraz niematerialnej w postaci porad prawnych czy psychologicznej. Analogicznie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do kolejnej z dyrektyw, której przepisy znajdują odzwierciedlenie w szeregu ustaw, w tym we wspomnianym Kodeksie karnym w zakresie dotyczącym przestępstw na tle seksualnym czy w Kodeksie postępowania karnego w odniesieniu do praw pokrzywdzonych dzieci, w tym co do szczególnego trybu przesłuchania, nagrywania takich przesłuchań, a także w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizującej również zapisy konwencji antyprzemocowej. Wiele z obecnie obowiązujących w naszym kraju przepisów, w tym również te jakże niezbędne z perspektywy osób pokrzywdzonych, te gwarantowane dziś prawem uprawnienia, które mogą się wydawać czymś oczywistym i podstawowym, zyskaliśmy dzięki naszej dotychczasowej obecności w Unii Europejskiej, dzięki dostosowywaniu polskiego prawa do prawa unijnego. Dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej nie tylko nasza infrastruktura drogowa, kolejowa się poprawia, gminy zyskują dofinansowanie, rolnicy zyskują dopłaty, a szkoły zostają docieplone i rozbudowane.

To właśnie praworządność, to właśnie prawa człowieka, to - tak jak w tym przypadku - prawa osób pokrzywdzonych. Przedłożony projekt ustawy wprowadza punktowe zmiany obecnie obowiązujących przepisów. Proponowane przepisy zmierzają do poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych, w tym do ustanowienia zasady domniemania wieku pokrzywdzonego, tak by rozszerzyć stosowanie szczególnych standardów odnoszących się do pokrzywdzonych osób poniżej 18. roku życia na osoby, których wieku nie można ustalić - np. cudzoziemców, których tożsamość jest nieznana - zaś ich cechy fizyczne i psychiczne mogą świadczyć o tym, że są osobami niepełnoletnimi.

Ponieważ są to zmiany korzystne i działające na rzecz osób pokrzywdzonych, w tym szczególności tych najmłodszych, do 18. roku życia, klub Lewicy popiera niniejsze przedłożenie i będzie głosował za skierowaniem tego projektu do prac w komisji. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Krzysztofa Paszyka, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści. Wykonałem to genialnie, przyzna pan. Bardzo dziękuję, panie marszałku, za oddanie pełnej nazwy klubu parlamentarnego, który mam zaszczyt reprezentować. Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Chciałbym przedstawić stanowisko klubu Koalicja Polska wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, zawartego w druku sejmowym nr 732. Projekt ten doprecyzowuje i uściśla obowiązujące przepisy odnoszące się do gwarancji procesowych przysługujących pokrzywdzonym. Wprowadza regulacje chroniące małoletnie ofiary przestępstw zgodnie z zasadą, że organ przeprowadzający przesłuchanie powinien zawsze kierować się dobrem dziecka.

Po zmianach w przypadku wątpliwości co do wieku pokrzywdzonego trzeba będzie stosować wobec niego uprawnienia procesowe takie jak wobec małoletnich. Rozwiązania z projektu sankcjonują obowiązującą praktykę dotyczącą oceny indywidualnej dla pokrzywdzonego i wskazują na konieczność szczególnego traktowania ofiary w postępowaniu karnym. Indywidualna ocena ma uwzględniać np.: cechy osobowe pokrzywdzonego, rodzaj, charakter i okoliczności przestępstwa, rozmiar doznanej szkody, a także relację między pokrzywdzonym a sprawcą. Ocena ta powinna także uwzględniać opinie, obawy i potrzeby pokrzywdzonego. Dodać należy także niezwykle istotny element tego przedłożenia, jakim jest implementacja przepisów Unii Europejskiej.

Panie marszałku, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Krzysztof Bosak, koło Konfederacja. Zapraszam, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Przedłożony projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego jest implementacją dwóch dyrektyw Unii Europejskiej, inspirowany jest troską o ochronę dzieci przed nadużyciami seksualnymi, w szczególności mamy tu na myśli dyrektywę w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. Polski system prawny prezentuje już w tej chwili dość wysoki standard obchodzenia się z ofiarami tego typu przestępstw, jednak te przepisy, które proponuje Unia Europejska, nie wyglądają źle. Jest domniemanie w przypadku osób, których wieku nie da się ustalić, tego, by traktować je jako osoby małoletnie, a więc stosować wyższe standardy ochrony, większą delikatność wobec ofiar tego typu przestępstw, szczególnie jeżeli chodzi o ofiary, których tożsamość trudno ustalić, a więc może to dotyczyć sytuacji dzieci porwanych - dzieci czy młodzieży, bo gdy mówimy o problemie z ustaleniem wieku ofiar, to dotyczy to młodzieży młodszej czy młodzieży na granicy dorosłości i wieku właśnie młodzieńczego objętych specjalną ochroną prawną - wówczas mogą to być sytuacje międzynarodowego handlu ludźmi i jak najbardziej podniesienie standardu ochrony jest czymś, o co warto zadbać. To drobna zmiana techniczna w Kodeksie postępowania karnego, natomiast przy tej okazji warto przyjrzeć się, jak wygląda realizacja zapowiedzi partii rządzącej w obszarze ochrony osób będących właśnie ofiarami przestępstw pedofilskich. Pozwolę sobie tutaj zacytować. Na konwencji wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w Szczecinie 12 maja 2019 r. lider PiS-u Jarosław Kaczyński, nieobecny niestety na sali w tej chwili, mówił: Chcemy w tych sprawach być naprawdę surowi, bezlitośnie surowi. Ani wysoka ranga w jakiejkolwiek organizacji, także kościelnej, ani nawet nagroda Nobla, ani nic innego nie zwalnia z odpowiedzialności w tego rodzaju sprawach. W konsekwencji w czerwcu 2019 r. partia rządząca przedłożyła w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu karnego zakładający m.in., że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat. Najbardziej zaburzonym sprawcom będzie grozić bezwzględne dożywocie, najcięższe zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać. Przypomnijmy, co się stało. W chaosie legislacyjnym projekt był przez Sejm przeprowadzony w sposób nieprawidłowy, niezwykle pospieszny, przez co nieprawidłowy. Prezydent Andrzej Duda wobec poważnych wątpliwości, czy projekt został w Sejmie uchwalony prawidłowo, skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny 14 lipca br. w wyroku sygnowanym KP 1/19 uznał, że ustawa jest niezgodna z konstytucją nie ze względu na swoją treść, ale ze względu na partactwo legislacyjne, które tutaj, w Izbie, się odbyło, i ten projekt trafił do legislacyjnego śmietnika, nigdy nie wszedł w życie. Partia rządząca nie przedstawiła ponownie tych przepisów w celu ich uchwalenia w Sejmie, a opinia publiczna o sprawie zapomniała. Pozwolę sobie też przypomnieć, że tak samo wiele miesięcy czekaliśmy na powołanie członków państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii i prace tej komisji w tej chwili właściwie dopiero ruszają, po tak długim czasie dyskusji na ten temat, organu, którego powołanie należy pochwalić, ale który zaczyna pracować w rok po tym, jak przepisy dotyczące jego stworzenia były w Izbie uchwalane. Oprócz prewencji oraz bezwzględnego ścigania przestępstw pedofilskich wobec małoletnich warto pochylić się też nad problemami opieki nad ofiarami. Stan ogólny psychiatrii dziecięcej w Polsce, jak już wszyscy wiemy w wyniku toczącej się debaty, jest opłakany. Dzieci z traumami wynikającymi z nadużyć seksualnych, z przestępstw i ze zbrodni o charakterze pedofilskim następnie nie mają dostępu do dobrej opieki, do dobrej terapii, która pozwoliłaby im wyjść z tej traumy. To jest też problem, który tutaj w Sejmie powinien być poruszony i powinien wybrzmieć. Poza takimi kosmetycznymi zmianami prawa wynikającymi z implementacji przepisów unijnych jak dzisiaj potrzebujemy też dotknąć tematu zbyt szybkiego, zbyt łatwego przedawniania się przestępstw pedofilskich oraz zbyt łatwej drogi do uniknięcia kary za ukrywanie takich przestępstw. Potrzeba tutaj znacznie bardziej kompleksowych zmian legislacyjnych. Partia rządząca takie zmiany zapowiadała, niestety one przepadły, nikt o tym (Dzwonek) w tej chwili nie pamięta. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Przechodzimy do zadawania pytań. Pierwsze pytanie zadaje pani poseł Joanna Fabisiak z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ustawa ma poprawić sytuację pokrzywdzonego. Ta ustawa jest potrzebna i jest dobra. Moje wątpliwości budzi jednak fakt przesłuchania i proszę o odpowiedź konkretnie na pytanie, czy prokuratorzy. Dotychczas prokuratorzy nie odbywają specjalnej specjalizacji, zatem możliwa jest sytuacja, że rano prokurator będzie prowadził dochodzenie w sprawie zbrodni, w południe w sprawie gospodarczej, a po południu będzie przesłuchiwał pokrzywdzone dziecko. Niezmierna wrażliwość takiego przesłuchania wymaga z całą pewnością przygotowania osoby, która będzie je przeprowadzała. Obecnie nie są i mówią mi to matki, które z takim problemem się zmagają. A zatem czy będą, czy też ta ustawa będzie tylko teoretyczna? Dziękuję bardzo. Dziękuję pani serdecznie. Pan poseł Wiesław Buż, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Celem jest wprowadzenie zmian do Kodeksu postępowania karnego zmierzających do uściślenia i doprecyzowania obowiązujących przepisów odnoszących się do gwarancji procesowych przysługujących pokrzywdzonemu. Wszystko jest okej, o czym tutaj pan minister mówił, kiedy wspomniał, jakie jest uzasadnienie projektu ustawy. Tylko dwa pytania. Dlaczego wobec tego te zmiany wprowadzamy po 8 latach od przyjęcia dyrektywy? Ile osób małoletnich narażono w ten sposób na ułomne postępowanie w tym czasie? Bardzo miło mi będzie usłyszeć od pana ministra kilka słów wyjaśnienia w tej sprawie, pana ministra, zresztą ziomka. Dziękuję bardzo. Przed nami sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan minister Marcin Warchoł. Dziękuję bardzo. Rozpocznę, panie marszałku, Wysoka Izbo, od drugiego pytania. Te dyrektywy implementował rząd Platformy Obywatelskiej, więc to pytanie jest do dzisiejszej opozycji. Dlaczego niepełna implementacja? Stan prawny w naszym kraju jest rzeczywiście taki, że mamy bardzo wysokie standardy ochrony praw pokrzywdzonych, ale one jeszcze nie wystarczają. Te dodatkowe przepisy, które proponujemy, mają ten standard jeszcze bardziej podnieść. Przechodzę do pierwszego pytania. Przecież to sąd przesłuchuje małoletniego pokrzywdzonego w sprawie o określone kategorie przestępstw. Ma to się odbywać tylko raz w trakcie postępowania przygotowawczego, chyba że na jaw wyjdą szczególne nowe okoliczności lub też oskarżony nie miał w trakcie przesłuchania swojego obrońcy. Ma to na celu ochronę przed wtórną wiktymizacją, żeby takiego dziecka nie ciągnąć po raz kolejny przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, później do sądu, często po kilku latach, jak to dziecko przeżywa traumę, i to traumę nieraz na lata. Dlatego absolutnie konsekwentnie opowiadamy się za zwalczaniem przestępstw pedofilskich - tutaj zwracam się do pana posła Bosaka - oczywiście tak, a wyrazem tego jest Kodeks karny, o którym tutaj mówiliśmy rok temu. W tymże Kodeksie karnym absolutnie będą przez nas proponowane ponownie wyłączenie przedawnienia przestępstw pedofilskich czy szereg innych zaostrzeń prawa w tym zakresie. Ofiara, powiadam, zostaje z traumą na całe życie.

Tak że jest to realizowane. Przypomnę, że przestępstwa gospodarcze, VAT-owskie dzisiaj są ścigane przez prokuratury regionalne. To w tych prokuraturach są najbardziej wykwalifikowani prokuratorzy, dzięki czemu mamy takie sukcesy, Prokuratura Krajowa ma takie sukcesy.

Sprawy lichwy, sprawy mafii lekowych, sprawy dopalaczy - to są już dzisiaj specjalizacje. Myśmy te specjalizacje wprowadzili dzięki reformie pana ministra Zbigniewa Ziobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, zawarty w druku nr 732, do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Dziękuję bardzo.

Wznawiam obrady. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Nie mam możliwości sprawowania swojego mandatu.

Jesteśmy przy głosowaniach. Szanowna Pani Marszałek! Chciałem zgłosić wniosek formalny o to, aby zwołać trzy połączone komisje. Właściciele pensjonatów, hoteli, kwater prywatnych, w większości rodzinne firmy nie mają możliwości skorzystania z pomocy. To jest dzisiaj tragedia tysięcy polskich rodzin. Apeluję o to, aby zwołać trzy połączone komisje w celu przyznania pomocy finansowej branży, która dzisiaj umiera i prosi o pomoc. Pan doskonale o tym wie. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 789 i 807) Proszę panią poseł Urszulę Rusecką o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zawarte w druku nr 807 o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 789. Marszałek Sejmu zgodnie z regulaminem Sejmu skierowała w dniu 30 listopada 2020 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia.

Wysoka Izbo! 47 tys. 47 tys. ludzi, którzy już nigdy nie zobaczą swoich dzieci, wnuków, rodziców. Do końca listopada w Polsce zmarło o 47 tys. więcej osób niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Do końca tego roku to będzie ponad 60 tys. zgonów więcej. I to osobiście obciąża pana, panie wicepremierze Kaczyński, bo to pan jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polaków. Chciałbym, żeby te liczby śniły się panu po nocach. Chciałbym, żeby wreszcie zrozumiał pan, że igranie bezpieczeństwem Polaków to zdrada stanu. Mieliście czas na to, by przygotować Polskę do drugiej fali pandemii. Zamiast tego pan, panie wicepremierze, wybrał partyjne gierki. Przecież miało nie być... ...wybrał pan przepychanki, walkę o stołki, zamiast doposażyć szpitale, zamiast wynagradzać medyków, zamiast zająć się tym, do czego powołani są odpowiedzialni politycy. Na pana sumieniu ciążą również tysiące zwalnianych polskich pracowników, tysiące zamykanych firm, bo zamiast pomagać przedsiębiorcom, zajmowaliście się sami sobą. I wreszcie, panie wicepremierze odpowiedzialny za bezpieczeństwo, od 6 października tego roku jedyną osobą, której poprawiło się bezpieczeństwo, to jest pan sam. To są dziesiątki radiowozów strzegących pana miejsca zamieszkania, tysiące policjantów ściąganych z całej Polski tylko dlatego, żeby zapewnić panu psychiczny komfort. Wstyd. To jest pana osobisty wstyd. Żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od tych wszystkich zaniedbań, rozpętał pan w Polsce piekło kobiet. Uzależniony od pana pseudo-Trybunał Konstytucyjny wydał nieludzkie orzeczenie, orzeczenie, które godzi w godność i elementarne prawo kobiet. orzeczenie, które nakazuje heroizm ponad ludzką miarę. Ale dlaczego pan to zrobił? Otóż zrobił pan to tylko dlatego, że nie potrafiliście sobie poradzić z pandemią i kryzysem. Chciał pan przykryć własną niekompetencję i niekompetencję własnego obozu. A potem co? Pałowanie kobiet? Urządził pan sobie na ulicach Polski rekonstrukcję stanu wojennego. Nie chcę przypominać, kto 39 lat temu spał do południa.

Ale dziś już wiemy, że nawet to skłócanie było robione pod publiczkę, tylko po to, by ukryć waszą bezradność. Wiemy, że tygodnie szargania wizerunku Polski w Unii Europejskiej, niszczenia pozytywnego dorobku pokoleń było panu potrzebne po co? By teraz uzasadniać kompromis, który zaprezentuje niemiecka prezydencja, a został przywieziony tu, do Polski, przez waszego wysłannika, który równie dobrze mógłby być wysłannikiem Putina, czyli premiera Węgier. Wstyd, panie premierze. Mam nadzieję, że jutro wbrew tym wszystkim złym podpowiedziom pan premier Morawiecki podpisze się pod dobrym, europejskim budżetem, ale zszarganie opinii Polski niestety jeszcze przez lata będzie ciągnęło się za naszym krajem, bo raz zburzonego zaufania nie da się tak szybko odbudować. Pan osiągnął to wszystko kosztem tego, że opinia publiczna i nasi partnerzy w Unii Europejskiej uważają rząd Polski za awanturnika, wręcz rosyjskiego agenta w łonie Unii Europejskiej. Chcę pana poinformować, że ta opinia w sumie niewiele odbiega od tej, którą miliony Polaków mają o panu. Za to wszystko pan będzie rozliczony, ale pana czas się skończył. Pan o tym doskonale wie i wiedzą również politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy siedzą dzisiaj obok pana w sejmowych ławach. Ale oni często buntują się przeciwko panu, już nie tylko w prywatnych rozmowach z nami, ale jawnie. Dlaczego? Wie o tym pan premier Morawiecki, wie o tym minister sprawiedliwości, dlatego toczą tak zażartą walkę o schedę po panu. Ale rozumieją to również obywatele. 70% Polek i Polaków chce pana dymisji. Ale to jest koniec kreowanych przez pana podziałów, koniec epoki szukania wrogów. Pan kończy tę karierę polityczną jako postać groteskowa. Okazał się pan bowiem tym wszystkim, z czym obiecał pan walczyć. To pan stworzył prawdziwy układ, to pan stał się symbolem elit oderwanych od rzeczywistości, to pan uczynił Polskę słabą i odizolowaną, to pan prowadzi Polskę do ruiny.

Podeptał pan wartości, na których przed 20 laty zbudował pan z bratem polityczny projekt Prawa i Sprawiedliwości. Ale dość już o panu. Pora opowiedzieć o Polsce, której nie będzie już nam urządzał prezes PiS. Polacy obudzili się. To widać na każdym kroku. Widać na ulicach, widać w sieci. Do głosu doszły miliony obywatelek i obywateli, którzy chcą żyć w innym kraju, kraju tworzonym przez nich i dla nich, dla wszystkich. Oni chcą Polski opartej na współpracy, Polski jasnych procedur i silnych instytucji, rządu, który nie mnoży problemów, lecz je rozwiązuje. I wam, którzy w tej chwili protestujecie na ulicach, walcząc o swoje prawa, chcę jasno powiedzieć: dziękujemy, ale też przepraszamy. My też nie jesteśmy bez winy. Za długo pozwalaliśmy, by Jarosław Kaczyński wodził nas za nos, by cała polityka koncentrowała się wokół wyreżyserowanych przez niego awantur. Daliśmy sobie przyprawić gębę totalnej opozycji i anty-PiS-u. Pora z tym skończyć. Po ponad 5 latach niszczenia więzi społecznych, niszczenia relacji od poziomu rodziny aż po Europę. nam wszystkim należy się nowy projekt, projekt, który przywróci Polakom nadzieję. Musimy działać razem. Koalicja Obywatelska, Lewica, ludowcy, ruchy pozaparlamentarne, ale również część z was, polityków Zjednoczonej Prawicy, bo przecież dla wielu z was dobro Polski jest również najważniejsze. Teraz czujecie się zagubieni i bezsilni w tym festiwalu oskarżeń, zaniedbań i fanatyzmu. Szanowni Państwo! To wotum nieufności nie jest przeciwko wam. Wręcz odwrotnie, bo tak samo jak my potrzebujecie dziś nowego otwarcia, dialogu i współpracy, bo Polskę uratować możemy tylko wspólnie. Przypomnijcie sobie wartości, dla których poszliście dla polityki.

Wysoki Sejmie! ust. 2 regulaminu Sejmu wniosek posłów opozycji, posłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, w sprawie wotum nieufności wobec wiceprezesa Rady Ministrów pana premiera Jarosława Kaczyńskiego skierowała do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która dzisiaj obradowała przez cały dzień, przez ponad 8 godzin, na dwóch posiedzeniach połączonych ze sobą tematycznie, intencjonalnie i emocjonalnie.

które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Polsce. komendanta głównego Policji, ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego.

A potem, na tym drugim posiedzeniu komisji właśnie, został zaprezentowany przez pana posła Adama Szłapkę wniosek w sprawie wotum nieufności wobec pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, rozpisany później na głosy wielu posłów opozycji. Większość członków komisji uznała, że wniosek jest bezzasadny, bezzasadny merytorycznie, [[Oklaski]] chybiony formalnie i politycznie i w głosowaniu zaopiniowała go negatywnie. 20 głosów było za negatywną opinią, 14 za pozytywną opinią wniosku. Pan poseł Adam Szłapka z nie mniejszą dawką nienawiści politycznej, niż teraz to zrobił pan przewodniczący klubu. zaprezentował ten wniosek. On obfitował w obraźliwe sformułowania, kłamstwa, obfitował w inwektywy. Ja musiałem zaprotestować przeciwko temu, odbyła się pewna polemika, ale właśnie tak to jest, proszę państwa. Mieliśmy wrażenie, że tym wnioskiem, wnioskiem o wotum nieufności dla pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, chcecie odreagować swoje frustracje. swoje przegrane wybory, to, że nie możecie wrócić do władzy, bo społeczeństwo was nie chce.

Można powiedzieć także, że przypisaliście mu 10 plag egipskich. Ale, szanowni państwo, nie załatwicie wnioskiem o wotum nieufności tego, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, a nie wy. Społeczeństwo wam dawno podziękowało.

Ta dyskusja nic nie dała, była bardzo emocjonalna. Wy pozostaliście przy swoich inwektywach, obraźliwych sformułowaniach, kłamstwach, bezpodstawnych zarzutach. Jeszcze raz, powtarzam: komisja zaopiniowała wniosek negatywnie i nie mogła postąpić inaczej, bo wniosek jest bezzasadny, bezsensowny, bulwersujący i ze wszech miar chybiony.

Otwieram dyskusję.

Nie są dopuszczalne pytania jako odrębny element debaty.

Panie Premierze! Wysoka Izbo! Pandemia COVID-19 zmieniła całe nasze życie, zmieniła cały świat. działania opozycji w Polsce. Zgłoszony przez państwa wniosek jest całkowicie bezzasadny, niemerytoryczny i niepoważny. Ten wniosek całkowicie nie ma sensu. Nie macie nic do zaproponowania poza atakiem. Gdy pan prezes Jarosław Kaczyński miał zostać wicepremierem, jeszcze zanim odebrał oficjalnie nominację, wy już chcieliście go odwołać, tak dla zasady, nieważne za co, byle by tylko była polityczna awantura. To najlepiej pokazuje, czym w istocie jest ten wniosek. Nic się nie zmieniliście, jesteście nadal totalną opozycją bez pomysłu, bez woli wsparcia państwa. z jedynym programem odsunięcia PiS od władzy. W waszym wniosku nazwisko Kaczyński pada blisko 50 razy. To jest najlepsze podsumowanie, o co w tym wszystkim chodzi. My zajmujemy się sprawami Polaków, rozwiązujemy ich problemy. Wy niezmiennie zajmujecie się prezesem Jarosławem Kaczyńskim oraz Prawem i Sprawiedliwością.

Ciężar działania poszczególnych resortów spoczywa na konkretnych ministrach, a funkcja, którą pełni pan prezes Kaczyński w rządzie, jest potrzebna, by była należna koordynacja i współpraca. To spójne i sprawne działanie jest dziś bardzo potrzebne, jest potrzebne jak nigdy wcześniej i daje konkretne efekty. Dziś wszystkie służby współpracują, współdziałają i wspierają się w działaniach, szczególnie w tym specyficznym czasie, czasie pandemii. Mówiąc o bezpieczeństwie, warto przypomnieć to, co się działo w roku 2015 i wspomnieć o działaniach pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w tym czasie. To właśnie wtedy pan prezes Jarosław Kaczyński jako pierwszy miał odwagę sprzeciwić się przymusowej relokacji migrantów, na którą zgodziła się ówczesna Platforma Obywatelska. Pamiętamy te słowa, te zapewnienia liderów Platformy Obywatelskiej: przyjmiemy każdą ilość. To właśnie pan prezes Jarosław Kaczyński na tej sali przestrzegał przed negatywnymi skutkami takiego działania. Dziś widzimy, kto miał rację. Ale ileż wtedy było ataków, ileż wtedy było nienawiści. Szanowni państwo, to właśnie pan prezes Jarosław Kaczyński uchronił Polskę przed takimi wydarzeniami, jakie widzieliśmy we Francji, jakie widzieliśmy w Niemczech, jakie widzieliśmy w innych krajach zachodniej Europy.

A co robiła Platforma Obywatelska? Wyśmiewaliście żołnierzy ochotników i całą formację. Nazywaliście ich wojskiem weekendowym. Mówiliście o tym, że to niemożliwe, żeby tym żołnierzom powierzyć cokolwiek poważnego. Jeżeli macie choć odrobinę honoru, to dziś powinniście przeprosić za tamte nikczemne ataki na całą formację Wojsk Obrony Terytorialnej. Plan bezpieczeństwa dla Polski, jaki wprowadza w życie pan prezes Jarosław Kaczyński i rząd Zjednoczonej Prawicy, to wymierne liczby i rzeczywiste działania. Podziwiam pracę polskich policjantów - bohaterów czasów pokoju. Dzięki ich ciężkiej i profesjonalnej pracy Polska jest bezpieczna, obywatele są bezpieczni. To właśnie dzięki takiej polityce naszego lidera Jarosława Kaczyńskiego zdecydowana większość obywateli czuje się bezpiecznie. Równie wysokie było do niedawna zaufanie do Policji, ale niestety dziś to zaufanie jest przez was niszczone. Chciałbym to jasno powiedzieć, że ręka podniesiona na policjanta to ręka podniesiona na polskie państwo i wy braliście w tym nikczemnym ataku udział. Jest mi za was wstyd. Na przestrzeni ostatnich lat Policja każdą taką manifestację ochraniała, bez względu na to, jakie były poglądy głoszone podczas takich manifestacji. Ale nie w czasie pandemii, bo to jest zagrożenie. Szanowni Państwo! Chciałbym podkreślić, że musicie się nauczyć, że wykonywanie mandatu posła nie polega na tamowaniu ruchu na ulicy. Żadna legitymacja nie zwalnia od przestrzegania prawa. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zaapelować do opozycji i powiedzieć jasno, że nie poprzemy tego wniosku. Ten wniosek jest całkowicie niezasadny, bezpodstawny. I moja rada: mniej o prezesie Jarosławie Kaczyńskim i o Prawie i Sprawiedliwości, a więcej o Polsce.

Wysoka Izbo! Bezpieczeństwo to stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania. Tyle w teorii. Bo praktyka pokazuje, że Jarosław Kaczyński postrzega je na opak. To pierwszy w historii cywilizowanych państw wicepremier do spraw bezpieczeństwa, który zajmuje się sianiem nienawiści, który chce, by obywatele żyli w atmosferze stanu wojennego, który w czasie pandemii wznieca protesty i, podgrzewając emocje, sprawia, że brutalizują się działania Policji. Policji, która doczekała się olbrzymiego kryzysu społecznego zaufania.

Pałka w ręku policjanta to obciążający Jarosław Kaczyńskiego symbol, wyraz odwetu na narodzie, którego nie rozumie i nie szanuje. Takie zachowanie przywodzi na myśl znane z historii szaleństwo władzy: władzy, która realizowała psychopatyczne rozkazy, niszcząc kraj, społeczeństwo i demokrację, władzy, której upadający reżim podnosił rękę na obywateli, podnosił rękę na kobiety. Tak wygląda strach Kaczyńskiego, strach przed kobietami, strach przed obywatelami, strach przed całym społeczeństwem. Bezpieczeństwo to też bezpieczeństwo zdrowotne. Bez strategii walki z pandemią dziś służba zdrowia pogrążona jest w chaosie, bez kadr i potrzebnego dofinansowania. Kiedy szpitale powiatowe walczą o przetrwanie, władza topi miliony w Szpitalu Narodowym, który zamiast pacjentami wypełniony jest propagandą. Bezpieczeństwa przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w pandemii, też Jarosław Kaczyński nie zbudował. Wiele branż nie przetrwa, wiele branż upadnie. Jarosław Kaczyński jest autorem polityki konfliktowania Polski z Europą. Z premierem Węgier sympatyzującym z Putinem realizują rosyjską strategię rozbijania Unii Europejskiej. To wszystko jest zaprzeczeniem bezpieczeństwa. To przerażający rekord. W 2 miesiące ostatecznie skonfliktował pan Polaków, wyprowadził Polki na ulicę i pogrzebał resztki relacji Polski z Unią Europejską. To hańba dla Polski, że ktoś tak nienawidzący Polki i Polaków jest w rządzie. To hańba dla Polski, że ktoś taki zajmuje się bezpieczeństwem Polaków. Jarosław Kaczyński stracił panowanie już nad wszystkim. Nie panuje nawet nad swoimi własnymi emocjami. To zachowanie musi zostać ocenione nie tylko politycznie. Tę ocenę wystawiamy, zgłaszając wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera Kaczyńskiego - człowieka, który na wielką skalę szczuje Polaków przeciwko sobie. Strach daje się we znaki wicepremierowi, który krzyczy, że będziemy siedzieć, bo sam boi się więzienia. Krzyczy, że mamy krew na rękach, by wyprzeć własną winę wobec narodu. Poprzez wotum zwracamy się do posłów PiS: odwagi, dajcie znać swojemu liderowi, że nie panuje już absolutnie nad niczym, a to zagraża życiu i zdrowiu Polek i Polaków. Pamiętajcie, wasza zgoda jest waszą współodpowiedzialnością. I na końcu - panie Jarosławie Kaczyński, depcząc praworządność, zbudował pan pełną podziałów, nienawiści, ideologii i propagandy Polskę. Za wszystko pan odpowie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Pan premier Kaczyński powiedział kiedyś, że chciałby być emerytowanym zbawcą narodu. Dziś rzeczywistość zweryfikowała pańskie słowa. Odkąd został pan wicepremierem, od października, odbyło się ponad 3,5 tys. protestów przeciwko pana rządom. Czy wtedy, 26 lat temu, chciał pan Polski podzielonej na lepszy i gorszy sort? Czy chciał pan Polski, w której politycy pod rękę z Kościołem chcą torturować kobiety? Czy chciał pan kraju, w którym mieszkańcy pozbawieni są niezawisłego sądu, sędziowie szykanowani, a superprokurator kryje Czy chciał pan Polski, w której Sejm jest atrapą, maszynką do głosowania? Czy chciał pan Polski zasnutej smogiem i wypalonej pożarami?

Panie Premierze! Odważny polityk staje przed komisją, w której jest procedowany wniosek o odwołanie. A dzisiaj panu premierowi tej odwagi zabrakło. Pamiętam, jak kilka miesięcy temu prezes Kaczyński wchodził do rządu, aby być jego stabilizatorem w czasie kryzysu i pandemii. Prawda jest jednak taka, że został pan wicepremierem, żeby walczyć z układem, ale we własnym rządzie. Miał pan łagodzić spory, tyle że między własnymi ministrami. Chciał pan nadzorować prokuratora generalnego, ale po to aby nie zamykał w więzieniu pańskich kolegów. I w końcu pan premier ma dbać o interesy własnych ludzi, którzy robią te interesy na maseczkach, respiratorach czy szczepionkach. Pan miał odpowiadać za bezpieczeństwo i odpowiada pan, tyle że za spokój swoich partyjnych koleżanek i kolegów. Skoro jest inaczej, niż mówię, panie premierze, to co pan premier naprawił w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy? Czy skończyło się ręczne sterowanie prokuraturą, rozsyłanie listów z instrukcjami, kogo wsadzać do więzienia, kogo nie, unikanie śledztw w sprawie księży pedofilów, inwigilacja opozycji i księży, upolitycznienie mediów czy w końcu umarzanie śledztw przeciwko swoim? Myślicie państwo, że jesteście blisko ludzi, ale wy tylko tak mówicie, bo jesteście dzisiaj elitą, która ma gdzieś zwykłych ludzi. Premier od bezpieczeństwa, zamiast uporządkować służby czy prokuraturę, zajmować się walką z pandemią, wspierać medyków czy tworzyć plan ratunkowy dla gospodarki, zarządza ze swojego centrum PiS-owskiego wszechświata na Nowogrodzkiej i namawia współpracowników, aby wetowali unijny budżet. Wicepremier Kaczyński miał być jak szeryf, niczym postrach z filmów o Dzikim Zachodzie. Okazał się pan jednak marnym stróżem prawa, a Dziki Zachód zafundował pan Polkom walczącym o swoje prawa. 22 października pan Kaczyński wydaje rozkaz swojemu osobistemu Trybunałowi Konstytucyjnemu, żeby dokonał barbarzyńskiego zamachu na prawa kobiet. 5 dni później, 27 października, pan Kaczyński, zirytowany protestami, wygłasza swoje orędzie, wzywa do przemocy. Na efekty nie trzeba długo czekać. Kilka godzin później 64-letni mężczyzna w Gdyni atakuje grupę młodych ludzi, wyzywa i wykrzykuje polityczne hasła, w końcu nożem rozcina twarz 23-latkowi. W następnych dniach grupy zamaskowanych sprawców napadają na protestujących we Wrocławiu, w Białymstoku i Warszawie. Kiedy protesty w obronie praw kobiet się nasilają, zamyka się pan premier w domu i otacza kordonem tysięcy policjantów. Zamiast kroku wstecz postanawia pan dokręcić śrubę. Do tłumienia protestów wysyła pan uzbrojone po zęby oddziały policyjne, które często mają charakter antyterrorystyczny. Prokuratura nakazuje ścigać i nękać organizatorów protestów. W Sejmie z mównicy wykrzykuje pan, że opozycja ma krew na rękach. Gdy alarmujemy, że policja zatrzymała posła Kopca, posłankę Falej, Kucharską-Dziedzic, wicemarszałka Czarzastego, pan się uśmiecha. Kiedy pryskają gazem w twarze posłanki Biejat i Nowackiej, pan mówi: Im się należało. Znalazł pan wroga w nowym pokoleniu. To jest właśnie tablica, która ma to pokazać. To w nim pan dostrzega. Młodzi.

Za to ma pan pełny plecak nienawiści. Symbolem pana rządów i drugiej kadencji PiS-u jest pałka teleskopowa. Kto nie umie ponosić odpowiedzialności, nie powinien pełnić państwowych funkcji. Jarosław Kaczyński dziś jest kłębkiem nerwów. Targa nim gniew i chęć zemsty. Jarosław Kaczyński, zamiast budować bezpieczeństwo, jest dziś architektem przemocy. Czas przerwać ten szaleńczy taniec. Dlatego Lewica zagłosuje za tym, żeby pan zakończył swoją misję i przestał być wicepremierem polskiego rządu. Pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, Koalicja Polska - PSL. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Słuchać Polaków, zmieniać Polskę - to było kiedyś wasze hasło. Jak słuchacie Polaków, to wiemy - po liczbie protestów i grup społecznych, które w tych protestach uczestniczą, od rolników po przedsiębiorców, od kobiet po osoby niepełnosprawne. Domagaliście się, żeby dzisiaj w tej debacie było więcej o Polsce, to usłyszycie teraz prawdę o tym, jak tę Polskę w ostatnich latach zmieniliście - według zasady: dzielić i zawłaszczać. Podział i zawłaszczenie. Podział na lepszy i gorszy sort. Podział medyków, prawdziwych bohaterów współczesnej Polski, na tych, którym się należą dodatki, i tych, którym pieniądze tydzień temu odebraliście. Pracodawców i przedsiębiorców podzieliliście według PKD, a nie według wielkości strat, które ponoszą przez COVID, i nie daliście im wsparcia. Samorządowców wczoraj podzieliliście na tych, którzy mają PiS-owską legitymację i dostali pieniądze z funduszu inwestycji lokalnych, i tych, którzy tej legitymacji nie posiadają - i mieszkańcom tej wspólnoty obywatelskiej się nic nie należy. Podzieliliście dziennikarzy i media. Podzieliliście media na te, które są patriotyczne, i te, które są, przecież wiadomo, z ukrytej opcji. Podzieliliście nawet koła gospodyń wiejskich - na te, którym się należą dotacje, i te, które w ARiMR się nie zarejestrowały i którym dotacji nie dacie. Ale, co najgorsze, podzieliliście Polskę, podzieliliście nasz ukochany kraj. Podzieliliście w ten sposób, że nie ma gwarancji bezpieczeństwa, bo to nie liczba F-35 gwarantuje bezpieczeństwo, ale wspólnota Polaków, wspólnota narodowa, świadomy swoich praw i obowiązków naród. A wy ten naród, tę wspólnotę rozbiliście. Zawłaszczyliście instytucje państwowe, z których uczyniliście PiS-owski folwark, sądy, z których sprawiedliwość jest uciekinierką, media, które są waszą tubą propagandową. Dołożyliście teraz koncern naftowy, który ma być koncernem propagandowym. Zawłaszczacie historię, bo uznajecie, że ona się zaczyna w 2015 r. Ale, co najgorsze dla osób wierzących, dla wspólnoty chrześcijan, zawłaszczacie, próbujecie każdego dnia zawłaszczyć Kościół. Oprócz podziałów i zawłaszczenia jest jeszcze wyzysk i odrzucenie. Wyzysk tych, którzy na was zagłosowali, a których po wyborach odrzuciliście. Wyzysk rolników, którzy wam zaufali, a którym zafundowaliście likwidację i zaoranie polskiego rolnictwa. Wyzysk frankowiczów, którym nie pomogliście. Wyzysk pokrzywdzonych przez organy państwa, którym obiecaliście skargę nadzwyczajną, na którą czekają już prawie 1000 dni. Wyzysk przedsiębiorców, na których codziennie nakładacie nowe podatki, choćby w ostatnich tygodniach, podatek od spółek komandytowych, podatek cukrowy czy podatki, które uderzą ich w przyszłym roku. Słuchać Polaków, zmieniać Polskę. A kogo wy dzisiaj słuchacie w waszym rządzie? Słuchacie radykałów, którzy chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Należy odrzucić ten głos radykałów, odstawić ich na bok i słuchać Polaków, którzy chcą być w Unii Europejskiej, chcą być silnym narodem w Unii Europejskiej. Przed nami ogromne wyzwanie: pokonać COVID. To jest wyzwanie dla całej wspólnoty narodowej, dla wszystkich Polaków, dla wszystkich obywateli. Pokonać COVID i przywrócić normalność. Dlatego proponujemy nową umowę społeczną, opartą na wartościach prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna. Te wartości niezależnie od tego, czy są czerpane z wiary, czy z innych źródeł, mają być podstawą nowej umowy społecznej, umowy społecznej, która doceni ludzi ciężkiej pracy, umowy społecznej, która zagwarantuje, że w naszym kraju będzie się chciało żyć każdemu, że będzie tutaj możliwa normalność, przyzwoitość, szacunek dla każdego człowieka niezależnie od poglądów i światopoglądu, w kraju, w którym jest przewidywalność i jest prawda. Możemy doprowadzić do tego, tylko przywracając normalność, odsuwając od rządu radykałów, którzy nie są i nigdy nie będą dobrym rozwiązaniem dla Polski. Dlatego Koalicja Polska. mając zawsze na pierwszym miejscu dobro i pomyślność obywateli, będzie głosowała za tym wnioskiem. A wy się tak naprawdę nie oburzajcie. Poseł Robert Winnicki, koło Konfederacji. Wysoka Izbo! Kaczyński do dymisji, mówiłem o tym jako pierwszy z tej mównicy. Tak, tak, pan premier Jarosław Kaczyński do dymisji, tak, szanowni państwo. Oczywiście nie ze względu na uzasadnienie, które padło tutaj z ust pana Borysa Budki, czy z ust przedstawiciela Lewicy.

Nie, to nie dlatego Kaczyński do dymisji. Kaczyński do dymisji. Już dajcie sobie spokój z tą czołobitnością, naprawdę. Już dajcie sobie spokój z tą czołobitnością. od ataku na rolników, od ataku bezsensownym projektem, od wymiany ministra rolnictwa na biernego, miernego, ale wiernego. Nie tylko dlatego, że w momencie, kiedy pojawiły się lewicowe manifestacje, to Jarosław Kaczyński odpowiadał za bierność Policji wobec ataków na kościoły, na miejsca kultu, na pomniki. Nie tylko dlatego, że Jarosław Kaczyński odpowiada za brutalne działania policji, dokładnie, toczka w toczkę, jak z czasów Donalda Tuska podczas Marszu Niepodległości 11 listopada tego roku. Identyczne zachowanie, identyczne procedury. No tak mówicie. Tylko nie wiadomo, co jest gorsze. Nie wiadomo, co jest gorsze. Czy to, że jest to plan polityczny - właśnie podgrzewanie emocji, niech atakują kościoły, będzie się działo, odwrócimy uwagę od kryzysu gospodarczego, od kryzysu systemu ochrony zdrowia? Niech się dzieje, niech będzie gorąco na Marszu Niepodległości, bo ludzie nie będą widzieli, w jakim kryzysie jest państwo. Czy, jak twierdzicie, to, że Jarosław Kaczyński za to nie odpowiada?

Jest kontynuacją SLD, jest kontynuacją Platformy Obywatelskiej. Jeśli dzisiaj Jarosław Kaczyński jest słaby, to właśnie dlatego, że nie ma żadnej zmiany, że jest wielkim kontynuatorem, również na polu polityki zagranicznej. Również w tym, że dzisiaj negocjowany jest kompromis, tak jak 11 lat temu podczas negocjacji traktatu lizbońskiego, kompromis, który de facto ma być kolejnym krokiem do centralizacji Unii Europejskiej. Kolejny krok, który będzie niszczył polską suwerenność. Poseł Artur Dziambor, koło Konfederacji. Panie marszałku, ja bym na początek prosił, żeby pan czasem uciszał klub. Tych też. Tych też. Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Jak słuchałem posła Tułajewa, to dziwiłem się, że to jest debata nad wotum nieufności dla premiera Kaczyńskiego, a nie debata nad przyznaniem mu Pokojowej Nagrody Nobla. Gdy dzisiaj rozmawialiśmy tutaj o merytorycznych punktach, poruszaliśmy np. temat akcyzy na samochody albo rozmawialiśmy o stoczni w Świnoujściu, którą właśnie zabiliście, zwalniając kilkaset osób z pracy, to było na sali dwóch reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz jest cała elita. Priorytety. Piękne. Szanowny Panie Wicepremierze do Spraw Bezpieczeństwa! Jak to jest piastować najbardziej fikcyjne stanowisko w tym rządzie? Bo przecież wiemy doskonale, że jest to stanowisko fikcyjne. Wiemy doskonale, że odbyła się tzw. rekonstrukcja rządu. Ta rekonstrukcja rządu polegała na tym, że kilku ministrów stało się wiceministrami. Kilku innych wiceministrów stało się dyrektorami nowych urzędów, które stworzyliście. Zlikwidowaliście kilka ministerstw, ale w zamian za to postawiliście urzędy i tam się więcej zarabia, bo nie funkcjonuje tam ustawa ograniczająca zarobki dla polityków. Widzimy to przecież. Wiemy o tym doskonale, jak to wygląda. Jest pan w tym rządzie, na tym stanowisku tylko po to, żeby dbać o bezpieczeństwo Mateusza Morawieckiego, który nie radził sobie w wojnie ze Zbigniewem Ziobro, oraz jest pan od tego, żeby pilnować tego, co się dzieje w środku, i nawet to panu nie wychodzi, bo na arenie międzynarodowej mamy wielogłos. Minister Gowin coś powie, minister Ziobro coś powie, premier Morawiecki coś powie na zewnątrz, przynosząc nam wstyd. Panie Premierze! Nie daje pan rady nawet utrzymać swojego rządu. Czas zrezygnować z tego stanowiska. Dziękuję.

Bardzo proszę, pani poseł Hanna Gill-Piątek. Bez tej latarki, jak pani może. Pani niestety nie potrafi tego wyłączyć.

Wysoka Izbo! Jego Ekscelencjo! Pana prywatne imperium, które pod przykrywką tzw. dobrej zmiany buduje pan przez ostatnie lata, trzeszczy w szwach. A pan dalej niby imperator rządzi i dzieli, a przydziela głównie swoim. To pana ludzie dokonali biznesowego rozbioru Polski. Ustalili nowe granice na mapie politycznej korupcji, tak aby nikt nie wchodził sobie w drogę. Za panem nie stoją już żadne idee. Żadne idee. W pana szeregach nie ma już oddanych dobru państwa działaczy opozycji demokratycznej. Pozostali Misiewicze, Szumowscy, nienawidzący kobiet ortodoksi z Ordo Iuris, wyszczekani chłopcy pana Zbigniewa Ziobry, miłośnicy serialu „Opowieść podręcznej”, jak np. pan minister Czarnek, córki leśniczych, biznesmeni importujący rosyjski węgiel, handlarze respiratorami oraz przy okazji bronią, sędziowie dublerzy, tajni współpracownicy służb PRL oraz konformistyczni zakonnicy Porozumienia Centrum. O bezpieczeństwo układu zamkniętego pana partii dba upolityczniona prokuratura, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będąca kpiną z prawa i skompromitowany Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Zawiadomienia o popełnieniu przestępstw słane do prokuratur przez obywateli i opozycję lądują w archiwach, bo na pana polecenie nadaje im się status makulatury. Niezliczonym urzędnikom, sędziom, funkcjonariuszom służb mundurowych pana pretorianie łamią kręgosłupy. Ogrom krzywd wywołanych przez pana politykę przeraża i przytłacza. To setki tysięcy ludzkich dramatów: policjantów, którym odebrano emerytury i dobre imię tylko dlatego, że kończyli edukację czy zaczęli służbę w czasach PRL. Kobiet i dzieci, traktowanych gazem na manifestacjach, włóczonych nocami po komisariatach czy nachodzonych po domach. Ale powiem panu słowami wiersza naszego noblisty: „Spisane będą czyny i rozmowy” Pamiętać to zszarganie państwa będą Polacy z pana pokolenia, dla których stał się pan symbolem zbrukania ideałów „Solidarności” Pamiętać też będą dzisiejsi dwudziesto- i trzydziestolatkowie. Te nowe pokolenia nie wierzą w paski TVP. Widzą za to pana czyny: plucie na konstytucję, zamach na prawo obywatelskie, nienawistne dzielenie rodzin przy wspólnym stole. Taki świat chce pan im zostawić. Perspektywa zdania władzy i rozliczeń budzi w panu lęk. Niesłusznie. Rewolucja „Solidarności” pokazała, że Polacy wiedzą, jak przywrócić krajowi wolność w sposób bezkrwawy i sprawiedliwy. Czy pamięta pan cokolwiek z tego? Bo chyba już nie. Dlatego, panie prezesie, czas na emeryturę. Chce tego aż 80% Polaków. Na emeryturę wysyłają pana wielkie miasta, małe miasteczka i wsie. Nawet w ocenie pana niedawnych zwolenników stał się pan nieznośnym wujkiem, który nie wie, kiedy wyjść z imprezy. Gdy 2 lata temu Polacy byli oburzeni sutymi nagrodami dla ministrów w rządzie Beaty Szydło, powiedział pan: Vox populi, vox Dei, głos ludu głosem Boga, i nakazał przeznaczenie nagród na cele charytatywne. Wtedy pan ludzi posłuchał. Dziś w imieniu 80% Polek i Polaków błagam, niech pan zejdzie ze sceny. Nie ma pan prawa ciągnąć nas za sobą do piekła, Polek i Polaków. Polska nie zasługuje na los, który chce nam pan zgotować. Zasługuje na lepszy rząd i lepszy parlament. Jedyną szansą uratowania Polski jest teraz przyjęcie uchwały o skróceniu kadencji Sejmu i jak najszybsze rozpisanie nowych wyborów. Pana czas minął i pan o tym dobrze wie. Tyle, że za 3 lata nasz kraj będzie dużo słabszy i dużo bardziej poraniony niż teraz. Niech pan ma tę przyzwoitość i skróci nam cierpienia. Być może słyszał pan kiedyś to zdanie: Tylko ci godni sprawować władzę, którzy mają dość siły ducha, by z niej zrezygnować. Ma pan dość siły ducha? Mając do wyboru siebie i Polskę, co pan wybierze?

Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta dobra strona, która teraz zabierała głos w tak zdecydowany sposób, w imię swoich powszechnie znanych i praktykowanych tutaj od lat demokratycznych przekonań - co prawda trochę kwestionowanych przez określenie ulica i zagranica, opozycja totalna - jednak pozwoli mi kilka słów powiedzieć. A zdecydują ci, którzy tutaj siedzą, i setki, tysiące innych z Prawa i Sprawiedliwości, ale także spośród wyborców. A kiedy będą wybory? No to wy lubicie czy lubiliście, bo już w tej chwili nie, lubiliście się odwoływać do konstytucji. Przemówienia, które tutaj słyszałem, były różne. Niektóre z nich zawierały pewną polityczną propozycję, cokolwiek przedwczesną i wskazującą na pewne niedoświadczenie tego, który tutaj w nieco bardziej cywilizowany sposób przemawiał. Cierpliwości, panie przewodniczący, cierpliwości. Ale ogromna większość tego, co zostało tutaj powiedziane, to jest pomieszanie absurdu, kłamstw, ale bardzo często też czegoś, co by można było określić jako projekcję własnych osobowości, własnej mentalności na kogoś innego. Rzeczywiście, jeśli wziąć pod uwagę waszą mentalność, wasze zachowania, wasz, powiedzmy sobie, bardzo głęboki brak kultury, to być może człowiek, który by jakoś personalizował. No ale, proszę państwa, my jesteśmy z zupełnie innego świata. Z zupełnie innego świata i wy najwyraźniej nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Nie jesteście w stanie zrozumieć tego, że ktoś naprawdę potrafi się kierować interesami Polski, [[Wesołość na sali]] a nie interesami swoich grupek. Tutaj padło jedno słowo rzeczywiście prawdziwe, chociaż w agresywnym przemówieniu. Otóż rzeczywiście z polskich sądów uciekła sprawiedliwość. Tylko to są wasze sądy. To pan Neumann mówił, co to za sądy. Bo ja jednak, i chciałbym tu młodego człowieka pouczyć, używam tej polskiej formy „pan” No być może pan już jest w innym kraju, tym na wschodzie. Tam się go rzeczywiście nie używa. To nie do pana Neumanna, tylko do innego młodego człowieka, który tutaj też przemawiał. No zastosowaliście też i taką socjotechnikę, która jest znana od wieków, od starożytności. Zmiana znaczenia słów i zmiana znaków wartości. Sięgnijmy do nieodległej historii. Nieodległej oczywiście w wymiarze historycznym, a nie w wymiarze ludzkiego życia. Związek Patriotów Polskich w istocie był agenturą NKWD zmierzającą do całkowitego zwasalizowania, podporządkowania, rozdeptania Polski. Następnie front demokratyczny czy obóz demokratyczny.

Panie pośle.

Zostały zastosowane także i przez was. Chociaż tych historycznych przykładów mógłbym tutaj bardzo wiele przytaczać.

odwoływanie się do tego, że ci, którzy są wzywani, mają broń.

Atakowanie kościołów to jest element pokojowych demonstracji, ale wzywanie do ich obrony to jest w gruncie rzeczy dzielenie narodu i wręcz przestępstwo. No tak, oczywiście, wzywanie do nienawiści - obrona kościołów przed różnego rodzaju aktami profanacji [[Wesołość na sali]] to jest wzywanie do nienawiści.

Być może także pana, panie pośle. Ale jeśli chodzi o prawdę, to prawda jest taka. że wyjątkowo wręcz wulgarne, niszczące polskie życie publiczne, można powiedzieć sprowadzające je na dno, wyjątkowo, jeszcze raz powtarzam, nieprzyzwoite pod każdym względem okrzyki i wypowiedzi, to wezwanie do dialogu. Otóż, szanowni państwo. Szanowni państwo, to jest właśnie wymiar tego zabiegu. Te czerwone litery, a właściwie cyfry, które tutaj widzę, zmuszają mnie niestety do skrócenia tego wystąpienia, a byłoby w tych sprawach jeszcze wiele do powiedzenia. Ale muszę jeszcze powiedzieć jedno. Jest instytucją koordynacyjną i zajmuje się problemami związanymi przede wszystkim z obroną narodową. Jeżeli chodzi o przyszłość, o to, co ma być uczynione, zrobione przygotowywanie zarówno rozwiązań prawnych, jak i praktycznych odnoszących się do tych dziedzin, mamy tutaj rzeczywiście, to przyznaję, dużo do zrobienia po bardzo, bardzo wielu latach różnego rodzaju zaniedbań. Ta praca zostanie wykonana. Wiem, wy będziecie się tym bardzo martwić, bo państwo będzie silniejsze, bo nie będzie już z tektury, już całkowicie nie będzie z tektury. To będzie w interesie Polski. Ale to będzie przeciwko opozycji totalnej.

To będzie po prostu Polska, gdzie będzie normalna - nie wiemy dzisiaj jaka, bo ludzie zdecydują, obywatele zdecydują - większość rządowa.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Opozycjo! Ten wasz wniosek, który skierowaliście przeciwko panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, to nie jest tak naprawdę wniosek o jego odwołanie jedynie, ale to jest próba zdezawuowania pewnej wizji Polski, którą prezes Jarosław Kaczyński proponuje. I dlatego chcę dzisiaj podczas mojego wystąpienia przed Wysoką Izbą przywołać kilka podstawowych różnic: wizja, którą proponował Jarosław Kaczyński wraz ze swoim bratem Lechem, versus wizja, którą proponowały tzw. elity III Rzeczypospolitej. Zacząć warto od tego, co było w ostatnim czasie tak bardzo widoczne: tyle państwa ataków na nas, tyle pytań, tyle frustracji, tyle oszczerstw, tyle kłamstw w kontekście COVID-19, ale ani razu nie padło jedno podstawowe pytanie z waszej strony: Jak możemy pomóc?

Niestety wasza postawa świadczy o tym, że nie tylko jesteście partią - zwłaszcza Platforma Obywatelska, opozycja - opozycją totalną, ale jesteście też opozycją zewnętrzną, partią zewnętrzną, partią zewnętrzną wobec polskich interesów, wobec polskiej racji stanu.

to wizja, która stawia polską rację stanu na pierwszym miejscu. A wasza wizja jest wizją bardzo wielu błędów, przeinaczeń, patologii i niedoskonałości w czasach III Rzeczypospolitej. I dlatego, szanowni państwo, warto zastanowić się nad przebiegiem ostatnich paru dziesięcioleci, bo premier Jarosław Kaczyński jest bez wątpienia, mogę powiedzieć, tą osobą, która na samym początku rozpoznała błędną, patologiczną naturę III Rzeczypospolitej i ją w bardzo konkretnych, bardzo precyzyjnych słowach obnażała.

To zaiste zupełnie odrębne wizje. Ale żeby to wszystko zidentyfikować, bo rzeczywiście zamęt pojęciowy, ta zapaść semantyczna.

I takie pytania Jarosław Kaczyński zadał. Na początku już pytał o to, na czym ma polegać realna demokracja, czy realna demokracja jest tylko pewnym rytuałem głosowania. przy nierównowadze sił społecznych, w którym po jednej stronie są media, jest władza. jest wsparcie Zachodu, a czasami Wschodu. i nie ma szans na realną zmianę władzy, jak to było przez praktycznie kilkanaście lat, czy realna demokracja ma polegać na oddaniu głosu narodowi w rzeczywisty sposób.

Dalej pan premier Jarosław Kaczyński pytał. na czym ma polegać sprawiedliwy system gospodarczy: czy na tym, że panuje klientelizm, który rzeczywiście jest sprytną metodą z jednej strony kooptacji, a z drugiej strony podporządkowywania sobie pewnych grup, korporacjonizm pewnych grup - widzimy to do dzisiaj w różnych grupach zawodowych, w tym znaczeniu używam tego słowa - czy ma być na zasadzie równowagi społecznej systemem gospodarczym dającym możliwe równe szanse każdemu. I premier Kaczyński odpowiadał: tak, to jest dla nas kierunek działania podstawowy, równe szanse dla każdego Polaka. Te wszystkie pytania, podstawowe pytania dla budowania właściwej wizji Polski padły z ust Jarosława Kaczyńskiego już bardzo szybko. Ale w waszym wniosku, szanowni państwo, odwołujecie się również do ostatnich lat i mówicie: chcemy rozliczyć premiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego za ostatnie 5 lat, bo za to odpowiada. Drodzy Rodacy!

Podaję dane od września 2020 r. versus wrzesień 2015 r. A w ciągu 4 lat, pierwszych 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, nastąpił wzrost realnych wynagrodzeń - 19,5%, przewyższał jakikolwiek wzrost wynagrodzeń w jakiejkolwiek wcześniejszej czterolatce czy wcześniejszej kadencji. Rzeczywiście straszne, horror. Zadłużenie zagraniczne. Zadłużenie zagraniczne spadło o 20%. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, która jest miernikiem naszej niezależności względem finansowania zagranicznego. To jest prawdziwa miara odzyskiwania niezależności w takich pokładach, o jakich wam się nie śniło wcześniej. Za to trzeba panu premierowi podziękować.

To są dane, szanowni państwo, jakich w poprzednich pięciolatkach nie uświadczylibyście.

Ale wizja Polski i strategia dla Polski pana premiera Jarosława Kaczyńskiego opierała się zawsze o sprawiedliwość, o prawo, o godność. I myślę, że to prawo pan premier rozumiał nie tylko jako prawo od strony formalnej, prawo, które ma być wykonywane w Polsce, ale również jako prawo rozumiane pozytywnie, prawo do czegoś, prawo do godnego życia, prawo do sprawiedliwego wyroku, prawo do rzeczywiście wolnych wyborów, do tego, żeby obywatele głosowali w realnych, demokratycznych wyborach. I to też jest coś, co głęboko wam nie pasowało. To jest coś, co było wbrew waszej krótkowzrocznej wizji, wizji, która na dobrą sprawę opierała się na ciepłej wodzie w kranie rzeczywiście, [[Oklaski]] na braku zaoferowania realnych korzyści dla szerokich rzesz społecznych. Ale właśnie popatrzmy na to od tej strony. Szanowni państwo, właśnie polityka społeczna została zmieniona w sposób fundamentalny i na zawsze ten wielki deficyt solidarności III Rzeczypospolitej przez premiera Jarosława Kaczyńskiego.

które spowodowały, że ci, którzy byli w III Rzeczypospolitej najsłabsi, odzyskali swoją godność [[Oklaski]] - bezrobotni, pracownicy, matki samotnie wychowujące dzieci. To były grupy, które były w dużym stopniu albo lekceważone, albo wręcz upośledzone. To premier Jarosław Kaczyński, kierując politykę społeczną w stronę tych szerokich rzesz społecznych, odbudował ich możliwości realizacji planów gospodarczych, ich aspiracje indywidualne i ich prawo do godności. Szanowni Państwo! Wtedy wy mówiliście, że to jest niemożliwe. One są gdzieś może zakopane. I to pan premier Jarosław Kaczyński miał rację.

Nie jest możliwe zrealizowanie naszych celów bez poddania się woli Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie, mamy naszą politykę, nie przyjmujemy uchodźców. Okazało się, że Unia Europejska też przyznaje mu dzisiaj rację.

Jak bardzo myliliście się w czymś, co dzisiaj często już nawet w publicystyce oddanych wam bez reszty mediów nazywane jest mitami. Mitem takim, że kapitał nie ma narodowości - premier Jarosław Kaczyński mówił o tym od dawna - mitem takim, że państwo jest wrogiem ludzi, państwo jest czymś złym, państwo powinno być nocnym stróżem. To było po to, żeby różne grupy interesów w ramach właśnie klientelizmu realizowały swoje interesy (Gwar na sali), żeby uprzywilejowane grupy interesów mogły de facto pasożytować w dużym stopniu na reszcie społeczeństwa.

Podobnie w odniesieniu do handlu, w odniesieniu do kapitału, swobodnej cyrkulacji kapitału czy do podatków, które miały być tym czymś najgorszym, czymś złym. I chcę państwu powiedzieć też jako były minister finansów, że to właśnie dzięki prezesowi i jego determinacji mamy dzisiaj finanse publiczne.

że zrobiliśmy jednocześnie wielkie programy inwestycyjne. Doprowadziliśmy do tego, że dziesiątki miliardów złotych przeznaczamy na inwestycje.

W waszych czasach, kiedy kryzys był dużo mniejszy, mówiliście: jesteśmy odporni na wezwania ze strony przedsiębiorców, na ratowanie miejsc pracy, na ratowanie gospodarki.

na początku pandemii postawił przed rządem jako szef, lider obozu.

Widzieliście je państwo?

Budżet państwa polskiego jest w stanie. bardzo dobrym, w tak dobrym stanie, że w czasie pandemii COVID możemy realizować programy inwestycyjne. To jest determinacja i długotrwały efekt realizacji planów strategicznych pana premiera Jarosława Kaczyńskiego.

Znacie, pewnie część z państwa zna rodowody niepokornych. Inteligencja zawsze była po to, żeby służyć wspólnocie, żeby być ze słabszymi. To była rola inteligencji, tych niepokornych, tamtych niepokornych opisywanych przez Cywińskiego. tych wszystkich postaci literackich, jak dr Judym, Siłaczka czy latarnik Skawiński, ale także wielkich postaci naszej historii, które były tam wtedy opisywane, jak Limanowski, jak Rodziewiczówna czy Przesmycki.

Niestety inteligencja, która zaczęła się kształtować, tak to nazwijmy, w czasach III Rzeczypospolitej, zrosła się z salonem, stworzyła salon - nie wiem, jak to powiedzieć - była de facto częścią elity, pseudoelity.

polityki, a w ślad za tym - los społeczeństwa i dzięki temu - siłę Polski.

To jest wasza wina. Ale też chcę powiedzieć, że posługiwaliście się bardzo często taką pałką propagandową. Tymczasem zobaczcie, co teraz działo się w waszych szeregach, co niejako z waszych szeregów wychodziło: wandalizm, agresja, obrażanie ludzi, skrajna wulgarność i jeszcze raz ataki na Kościół.

To jest coś zupełnie odwrotnego do tego, jaką wizję, jaką propozycję dla Polski ma prezes Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo!

Słowo, liczy się słowo, to, żeby dyskurs opierał się o fakty, o to, co rzeczywiście nurtuje ludzi. I pan prezes Jarosław Kaczyński rzeczywiście nazwał we właściwy sposób zjawiska, które zostały przez was. Cały czas jest próba ich przeinaczania. Mówiliście bardzo często, że to leniwi ludzie, że to gnuśność, że mamy tutaj do czynienia, no, niestety z lenistwem. Rolnik jest też leniwy - to z waszej strony padało coś takiego - dlatego mało zarabia. Naród to pojęcie. Oj, uwaga, bo ono ociera się o nacjonalizm. Dzisiaj rzeczywiście cały czas domagamy się tego, co na początku, po transformacji nazwano dekomunizacją. Dzisiaj należy mówić o depostkomunizacji. Tak, cały czas to jest potrzebne. bo wy jesteście często fundamentem tego systemu. A więc granice naszego języka są granicami naszego świata. I dlatego wyznaczenie tych granic we właściwy sposób, określenie tych zjawisk przez prezesa miało fundamentalne znaczenie dla sformułowania potem oferty politycznej i oferty programowej. Panie Premierze! Słyszałem, że nasza tutaj szanowna opozycja ma pewien plan opracowania swoich idei. które ma zaprezentować w najbliższym czasie w formie, jak rozumiem, jakiegoś programu. No, serio? To ciekawe, że teraz wpadli na coś takiego. Bardzo się cieszę z tego, ale ja wam powiem, dlaczego wychodzi z was taki kompleks. dlaczego wy próbujecie wszystko przykryć krzykiem, kłamstwem, kpiną i drwiną. Polskość dla was to nienormalność, a dla Jarosława Kaczyńskiego - według niego za Polskę trzeba dziękować. Dziękować.

Tak, tak, wasze 10 stron nie przykryje tych lat, które były latami walki o lepszą Polskę, walki o sprawiedliwą Polskę, o sprawiedliwą i silną Polskę. I dlatego to właśnie droga Jarosława Kaczyńskiego spowodowała, że dzisiaj żyjemy w normalniejszym kraju, w normalnym kraju.

Ale jego idee i jego czyny żyją wśród nas i razem z nami budują lepszą i sprawiedliwszą Polskę.

Dziękuję panu premierowi. Zamykam dyskusję. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań.

Wznawiam obrady. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu.

Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 826. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Kontynuujemy głosowanie nad poprawkami Senatu. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 211. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Nikt nie był za, przeciw - 447, 1 się wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 216. poprawki, zechce nacisnąć

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 217. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 218. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Łącznie z tą poprawką głosować będziemy nad 226. poprawką. Głosujemy.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

Głosujemy.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Łącznie z tą poprawką głosować będziemy nad 433. poprawką. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 225. i 433., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 229. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Głosowało 450 posłów. Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 295. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 296. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 431. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 434. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 437. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 438. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 439. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

Głosujemy.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 443. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. W 444. poprawce do art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Senat proponuje nowe brzmienie ust. 8.

4 - za, 450 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 445. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy.

Nikt nie był za, 453 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 447. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Głosujemy.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 449. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 450. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Nikt nie był za, 455 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego. Przypominam, że zgodnie z art. 159 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Przystępujemy do głosowania.

Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec wiceprezesa Rady Ministrów pana Jarosława Kaczyńskiego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 826) Prezydium Sejmu na podstawie art. 20 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 826, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 9 grudnia br. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą.

Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów chce się jeszcze zgłosić? Jeżeli nie, zamykam listę. Bardzo proszę. Nie ma pana posła. Pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska.

Wysoka Izbo!

Tak, szanowni państwo, stanowią własność Skarbu Państwa.

Natomiast, szanowni państwo, jest tak, że to Skarb Państwa, który powinien brać odpowiedzialność właśnie za tę zwierzynę w stanie wolnym, przerzucił całą odpowiedzialność na Polski Związek Łowiecki.

Będziemy mieli parki narodowe, nie będziemy mieli prowadzonej gospodarki łowieckiej, rolnicy będą mieli coraz większe straty. Do kogo wtedy pójdą rolnicy? Do Skarbu Państwa.

Po drugie, o to, żeby te koła łowieckie, które są zagrożone swoim funkcjonowaniem, można było uratować.

Dlatego też, panie premierze, panie ministrze, jeszcze raz apeluję o pilną tarczę osłonową dla rolników na odszkodowania (Dzwonek) i o pilne rozpoczęcie prac nad nowym Prawem łowieckim. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Wysoki Sejmie! Może pan premier wysłucha też mojego oświadczenia, bo jest bardzo ważne. Oświadczenie w sprawie dramatycznej sytuacji branży turystycznej. Kilka minut temu większość sejmowa odrzuciła poprawki Senatu w sprawie pomocy dla branży turystycznej, tj. hoteli, pensjonatów, gastronomii i innych usług. Przedsiębiorcy tej branży od 3 miesięcy nie prowadzą działalności i tym samym nie uzyskują żadnych przychodów. W jaki sposób mają zapłacić ZUS, kredyty bankowe, wynagrodzenia pracownikom, pokryć koszty stałe obiektu? Jak mają wywiązać się z zawartych umów z Polskim Funduszem Rozwoju, który nakłada na nich obowiązek utrzymania zatrudnienia co najmniej przez 1 rok? Takie same problemy mają przedsiębiorcy związani z turystyką, a więc usługi pralnicze, sprzątanie i inne. Im także grozi bankructwo. W turystyce pracuje ponad 1 mln osób, które wypracowują rocznie ok. 7% PKB. Czy można tak lekceważyć tę grupę przedsiębiorców i gminy górskie i podgórskie? Dlaczego rząd nie podejmuje rozmów z branżą turystyczną i nie próbuje znaleźć rozwiązania w sprawie częściowego odmrożenia działalności? Samorządy i przedsiębiorcy doskonale wiedzą, jak zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne turystów i mieszkańców i jednocześnie nie burzyć wszystkiego, co dookoła funkcjonuje, ale nikt ich nie słucha. Tymczasem Czesi już ogłosili otwarcie hoteli, gastronomii i wszelkich usług w sezonie zimowym, oczywiście z ograniczeniami, ale są czynne. Czy nam nie zależy na turystach i chcemy dobrowolnie zrezygnować z olbrzymich dochodów, jakie ta branża przynosi, i przekazać je Czechom? Jak to nazwać? W Karpaczu jest na to nazwa, ja nie będę jej tu w tej chwili powtarzać. A co z decyzją w sprawie ferii zimowych? Wszyscy czekają na ferie: rodzice, dzieci i cała branża turystyczna. Wybitni specjaliści medyczni w zakresie leczenia i ograniczania zachorowań, w tym prof. Simon, jednoznacznie mówią, że wydłużenie wyjazdów na ferie jest bardzo pożądane i bezpieczne. Osoby, które przeszły chorobę, mogą bez ograniczeń korzystać z wszelkich usług turystycznych. Takich ludzi są setki tysięcy w Polsce. Dlaczego nie bierze się pod uwagę tych opinii?